Dziękuję.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pragnę przedstawić poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Wysoka Izbo!

Ten projekt ustawy jest wyrazem autentycznej troski i naszego poselskiego obowiązku, wręcz imperatywem kategorycznym, w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków, bezgranicznego ratowania ich życia i zdrowia w tak trudnym i dramatycznym okresie pandemii koronawirusa. Natomiast fundamentem i osnową treści tego projektu ustawy jest naczelna zasada w lekarskim przyrzeczeniu Kodeksu etyki lekarskiej: Salus aegroti suprema lex esto - zdrowie każdego chorego jest najwyższym prawem. Wysoka Izbo! Współczesny świat zadrżał przed niewidzialnym, ale jakże groźnym i przebiegłym wrogiem, koronawirusem, który zaatakował ponownie ze zdwojoną siłą. Cały świat, Europa walczą. Ten dramatyczny okres pandemii COVID-19 to trudny i szczególny czas, zatem musimy podejmować też trudne i szczególne działania. Byłoby wprost idealnie, gdybyśmy w imię solidarności międzyludzkiej działali wspólnie i w jedności, zgodnie z aktualnym hasłem: Wszystkie ręce na pokład. Zatem podwyższamy do 200% wynagrodzenie zasadnicze wraz z pochodnymi dla osób skierowanych przez wojewodę do pracy związanej ze zwalczaniem COVID-19. Wprowadzamy klauzulę miłosiernego samarytanina, inaczej system no-fault, bez winy, czyli niekaranie za niezawinione błędy medyczne w sytuacji ratowania ludzkiego życia. Wprowadzamy prawo do zachowania 100-procentowego uposażenia w okresie zwolnienia od zajęć służbowych z powodu stwierdzenia zakażenia lub zachorowania, kwarantanny, izolacji lub izolacji domowej w przypadku funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz żołnierzy Wojska Polskiego. Wprowadzamy możliwość skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii pracowników podmiotów medycznych, osób wykonujących zawody medyczne oraz innych, np. studentów zawodów medycznych, doktorantów, ratowników medycznych, lekarzy, którzy są w trakcie stażu podyplomowego, albo lekarzy, którzy ukończyli staż, ale jeszcze nie zdali lekarskiego egzaminu końcowego. Wprowadzamy przepisy umożliwiające w trybie uproszczonym, ale też pod ścisłą kontrolą właściwych konsultantów, okręgowych izb lekarskich, pod nadzorem specjalistów, zatrudnianie na określony czas lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską - ale pod ścisłymi restrykcjami i po spełnieniu określonych w ustawie wymogów.

Wprowadzamy możliwość zawieszenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital w przypadku odmowy wykonania obowiązku albo polecenia lub nienależytego wykonania, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, wniesienia skargi do sądu administracyjnego oraz automatycznego wygaśnięcia zawieszenia po upływie 30 dni od dnia odwołania epidemii. Ujednolicamy i uszczelniamy sposób wystawiania zaświadczeń lekarskich. Do istniejącego zapisu w ustawie o izbach lekarskich, art. 83 ust. 1 pkt 7, o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu lekarzy dodajemy możliwość pozbawienia prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym; oczywiście najczęściej to będzie dotyczyć lekarzy zatrudnionych spoza Unii Europejskiej. Wydłużamy okres realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Powszechnie znana jest starożytna sentencja Seneki Młodszego: W trudnościach odwołuj się do rozumu. Liczne szeregi naszych współczesnych bohaterów w służbie zdrowia, głównie na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, mogą się powoli uszczuplać. Choroba, izolatoria, izolacja domowa, kwarantanna, a nawet zgon - to główne powody osłabienia tej linii. Co ważne, oni też mogą stać się pacjentami. Zatem w imię solidarności zawodowej, solidarności społecznej oraz w imię świętej sprawy, jaką jest życie i zdrowie każdego obywatela, mamy święty obowiązek jego ratowania. Dziś nie czas na waśnie i kłótnie polityczne, na czarnowidztwo. Jesteśmy silni i pokonamy wroga, ale jeśli będziemy razem, zwyciężymy szybciej i bez tylu ofiar. Jednocześnie jesteśmy otwarci na dalsze, na dobre i korzystne rozwiązania w przedłożonych propozycjach, projektach ustaw opozycji. Proszę pana posła Zdzisława Wolskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy z druku nr 684. Panie Marszałku! 10 kwietnia rozporządzeniem Rady Ministrów nałożono na nas obowiązek noszenia maseczek, zasłaniania ust i nosa. Wtedy, w kwietniu, sytuacja w społeczeństwie była inna. Pamiętamy, że społeczeństwo było wyjątkowo zdyscyplinowane. Wtedy bardzo mało było sytuacji nienoszenia maseczek, a już na pewno - nienoszenia demonstracyjnego. Ale sytuacja się zmieniła, również w wyniku tego, że najwyżsi przedstawiciele władz państwa, z panem prezydentem, premierem, a nawet ministrem zdrowia, zaczęli do tego podchodzić lekceważąco z powodów politycznych.

Wszyscy ludzie myślący, słuchający naukowców wiedzieli już wiosną, że do epidemii, i to na dużą skalę, dojdzie. Teraz, nie mając za bardzo możliwości ochrony pacjentów przed następstwami COVID-u - to będzie przedmiotem odrębnych dyskusji - chociaż się chrońmy. W związku z tym Lewica zaproponowała zmiany w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z roku 2008. Ale było denialistów wielu, którzy kwestionowali maseczki, bardzo aktywnych. Zaczęły się procesy, w których sądy, zgodnie z aktualną literą prawa, kary za nienoszenie maseczek uchylały. Również w sytuacji gdy w sklepie ekspedientka odmawiała obsługi pacjenta bez maseczki, okazywało się, że to ekspedientka była karana. Chcemy to zakończyć. Proponujemy w naszym projekcie ustawy, by dokonać zmiany w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, by jednoznacznie minister zdrowia zarządzał obowiązek noszenia maseczek, również np. kasków w przypadku motocyklistów, które tę rolę spełniają - to są szczegóły - w miejscach użyteczności publicznej, czyli w placówkach handlowych, w transporcie zbiorowym, w placówkach usługowych, w sektorze bankowym.

W paragrafie właśnie w tej ustawie będzie jednoznaczny zapis dotyczący tych, którzy nie przestrzegają wytycznych zarządzenia ministra zdrowia. Będą oni ponosili karę grzywny już w sposób jednoznaczny, nie do zakwestionowania przez ewentualne sądy. Proponujemy również dodać artykuł o tym, że nienoszenie maseczek może być uzasadnioną przyczyną odmowy sprzedaży lub odstąpienia od oferty w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, czyli mówię również o przypadkach medialnych, kiedy to ekspedientka ponosiła karę.

Dziękuję. Dziękuję. Proszę teraz pana posła Dariusza Klimczaka o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy z druku nr 685. Wysoka Izbo! Nadszedł czas, przyszedł moment, w którym przedstawiamy ważne ustawy dla życia Polaków, dla systemu ochrony zdrowia. Dobrze, że dzisiaj zaczynamy o nich rozmawiać, ale wszyscy wiemy, że to jest działanie spóźnione i tylko dlatego następuje, że mamy pożar w systemie ochrony zdrowia. Polskie Stronnictwo Ludowe i klub Koalicji Polskiej przedstawiły ustawę, o której dzisiaj mamy możliwość mówić, już w marcu. Złożyliśmy ją w kwietniu, bo wtedy była największa potrzeba wyjścia z inicjatywą dodatków do pensji dla wszystkich pracowników systemu ochrony zdrowia, ale także dla pracowników społecznych, którzy udzielają świadczeń medycznych, którzy pomagają osobom zakażonym i podejrzanym o zakażenie. Wystąpiliśmy z taką inicjatywą, dzisiaj rząd także wychodzi z podobną inicjatywą, ale bądźmy świadomi, dlaczego rząd wychodzi z tego typu działaniem. Ponieważ pojawił się problem. My zaproponowaliśmy nasze dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników systemu ochrony zdrowia i pracowników społecznych nie tylko po to, żeby dać im dodatkowe honorarium, ale także po to, by wynagrodzić im tę bardzo ciężką pracę w zawodzie strategicznym, także uhonorować ich pracę. To powinno odbyć się na samym początku epidemii, a nie dzisiaj, kiedy rząd próbuje ratować sytuację. Szanowni Państwo! Ale przecież my wiemy, że dobry Samarytanin nie brał pieniędzy za pomaganie drugiemu człowiekowi. Dzisiaj wiemy, że to jest zasłona dymna, próba wielkiej łapanki ludzi do pracy w szpitalach. Prawo i Sprawiedliwość myśli, że za pieniądze wszystko załatwi, że kupi lekarzy za pieniądze. Tu trzeba dużo więcej delikatności.

Przepisy nie mogą być chaotyczne, zaskakujące, wprowadzane w sposób niezrozumiały, bo dojdzie do tego, do czego doszło w Czechach, w sytuacji kiedy wyjdzie wasz minister i powie to, co powiedziała pani minister w Czechach. To ma ścisły związek z naszą ustawą, ponieważ nasza ustawa była wyprzedzająca, dalekowzroczna. Premier Morawiecki patrzy tylko pod nogi, nie patrzy daleko przed siebie, a tego się oczekuje od osoby pełniącej najważniejsze funkcje w państwie. Dzisiaj wprowadzacie regulacje dotyczące maseczek, po tym wielkim chaosie, po tym, co mówił były minister Szumowski, po tym, co mówił główny inspektor sanitarny, dzisiaj to regulujecie, ale dojdzie do tego, że kiedyś będziecie musieli napisać regulacje dotyczące zakazu skoku na główkę do pustego basenu, bo do tego dotrze polityka informacyjna w państwie.

Brakuje konsultacji z samorządami. Gdzie jest ta współpraca, o której zawsze mówiliście? Uważam, że za parę godzin powinien wyjść na tę mównicę pan premier Morawiecki i posypać głowę popiołem.

Dzisiaj jak na dłoni widać wszystkie zaniedbania w systemie ochrony zdrowia, mało tego, widoczny jest brak działań, których nie podjęliście w czasie wakacji. Przespaliście całe wakacje. Szpital narodowy. To, że będziecie mieli dodatkowych zastępców? Pamiętam, kiedy z tej mównicy mówiliśmy o systemowych zmianach w inspekcji sanitarnej. A co wy zrobiliście? To, że powiatowego inspektora nie będzie powoływał starosta, tylko rząd?

Nie tego oczekują Polacy. Proszę pana posła Jacka Protasa o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy z druku nr 686. Wysoka Izbo! Samorząd terytorialny w Polsce odgrywa ogromną, niepodważalną rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania państwa. Realizuje 2/3 inwestycji w sektorze publicznym, odpowiada za organizowanie ogromnej większości usług dla mieszkańców. Samorząd jest właścicielem ponad połowy polskich szpitali. Samorządy organizują, nadzorują funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych, zapewniają mieszkańcom transport publiczny, odpowiadają za gospodarkę odpadami, dostarczanie wody i odbiór ścieków. Mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo i ład publiczny. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie są szefami zespołów reagowania kryzysowego na terenie swoich samorządów, zapewniają zatem bezpieczeństwo obywateli podczas wszelkich zagrożeń życia lub zdrowia. Podczas pandemii koronawirusa w Polsce samorządy wzięły na siebie ogromną ilość obowiązków, które wynikają z ich zadań, ale także takich, które w tym trudnym czasie powinny wykonywać rząd i administracja publiczna, a ich nie wykonują z różnych powodów. Podjęcie tych działań wymaga ogromnego wysiłku finansowego, co w i tak trudnej sytuacji finansowej samorządów wygenerowało ogromne kłopoty ze spięciem budżetów. Wymaga to również sprawnych, szybkich i skutecznych działań organizacyjnych. Dużą i częstą przeszkodą w tym skutecznym działaniu jest konieczność stosowania przez samorządy terytorialne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wydłuża to w sposób często niebezpieczny procedury zakupu usług, sprzętu i wyposażenia niezbędnego natychmiast do działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Chodzi w szczególności o środki zabezpieczenia indywidualnego takie jak maseczki, płyny dezynfekujące, odzież ochronna, przyłbice, testy itp., a także o niezbędny sprzęt dla szpitali, innych placówek medycznych, instytucji publicznych, które muszą sprawnie funkcjonować i wykonywać swoje zadania w warunkach pandemii. Dlatego jako Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska przedkładamy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, druk nr 686, która przewiduje możliwość dokonywania zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych. Oczywiście to prawo będzie przysługiwało jednostkom samorządu terytorialnego pod warunkiem, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Dla zapewnienia przejrzystości i transparentności tego procesu, co bardzo ważne, proponujemy, by zamawiający w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia zamieścili w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę firmy bądź imię i nazwisko podmiotu, z którymi zawarli umowę na wykonanie tego zamówienia. Wejście w życie tej ustawy będzie miało na pewno pozytywne skutki społeczne, umożliwi samorządom szybkie reagowanie i działanie w sytuacjach zagrożenia życia bądź zdrowia. Wejście w życie tej ustawy nie będzie miało też żadnych skutków dla budżetu państwa.

Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy, a w zasadzie pakietu projektów ustaw, o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, tj. propozycji zawartej w druku nr 683, a także odnieść się pokrótce do pakietu ustaw zgłoszonych przez kluby opozycyjne.

Najważniejszą kwestią tej ustawy, którą całym sercem popieram, jest pewne uporządkowanie prawne i jednocześnie takie hasło, które dzisiaj, w sytuacji pewnego zaskoczenia, panie pośle, nikt na świecie nie przewidział, że druga fala epidemii będzie miała taki, a nie inny wymiar. Ona służy temu, żeby wszystkich możliwych pracowników ochrony zdrowia, którzy chcą być i którzy będą zaangażowani w proces zapobiegania, testowania, jak również leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, zwolnić z obowiązku odpowiadania za niezawinione błędy. Błąd lekarski jest istotą każdej pracy lekarza, on się zdarza na wielu różnych frontach, to jest błąd i osobisty, i leczniczy, ale to jest też błąd organizacyjny, wiele takich błędów znamy.

Mówimy również o tym, co jest w propozycji Koalicji Polskiej, żeby podnieść gratyfikację dla tych pracowników, którzy są i będą zatrudnieni w ramach walki z koronawirusem, i proponujemy podniesienie tej pensji o 200% wynagrodzenia zasadniczego. Oczywiście są co do tego przeprowadzone odpowiednie symulacje, ponieważ każda ustawa wymaga opisania skutków finansowych regulacji.

Przy czym jeżeli będzie 2%, 3%, 4%, to te szacunki wzrosną. Na dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, myślę, nikt na tej sali nie jest w stanie przewidzieć, ilu pracowników będzie zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Pragniemy również - to było już w poprzednich regulacjach - żeby jeżeli ktoś ulegnie zakażeniu albo będzie w jego przypadku konieczność kwarantanny, zasiłek z tego tytułu niezdolności do pracy był w wysokości 100%, a nie, jak dotychczas, 80%, bo jak państwo wiecie, ZUS wypłaca za pierwszy miesiąc niezdolności do pracy 80% podstawowego wynagrodzenia.

Wiemy, że z tym jest ogromny problem. I proszę państwa, to nie jest tak, że wszyscy, którzy dostaną skierowanie do pracy, zaraz będą musieli się stawić. Pierwsza sprawa to bezwzględnie współpraca z izbą lekarską, czyli z tymi, którzy posiadają pełne dossier pracownika ochrony zdrowia, jakim jest lekarz, i ta współpraca musi również (...) kwalifikacje.

Ale to jest oczywiście nieobligatoryjne. Ci lekarze również mogą pracować i to nie jako wolontariusze, ale jako pełnopłatni członkowie zespołów terapeutycznych. Chcieliśmy również zaprosić - to też już jest uregulowane w ustawach - lekarzy specjalistów z krajów spoza Unii Europejskich. Tutaj na okres pandemii zastosowaliśmy szczególne przepisy, oczywiście pod tymi samymi warunkami, jakie są w ustawie, nad którymi procedowaliśmy bodajże 2–3 miesiące temu. Już dzisiaj lekarze specjaliści spoza Unii Europejskiej mogą u nas pracować. Mówiliśmy również o tym, że jest bardzo ważne, żebyśmy rozwiązali problem tych lekarzy, którzy specjalizacji nie mają, ale mają określoną wiedzę medyczną, być może jeszcze nieugruntowaną albo nieukierunkowaną na choroby zakaźne. Chodzi o to, żeby oni również mogli pracować i żeby mogli również być zatrudnieni.

Inne uregulowania dotyczą raczej spraw związanych z częścią organizacyjną. Przede wszystkim będzie powołany zespół wsparcia Państwowego Ratownictwa Medycznego. To bardzo ważne.

Na koniec powiem, że oczywiście cieszę się z jednego faktu - to tu nie wybrzmiało w tych ustawach - że przy premierze powstał wreszcie zespół składający się z fachowców: epidemiologów, wirusologów, który będzie starał się wypracować jedną linię informacyjną.

Bardzo dziękuję, panie pośle. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska pan poseł Cezary Tomczyk. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Myślę, że wszyscy powinniśmy korzystać z tego doświadczenia, bo widzimy, że przepisy przygotowywane na kolanie są po prostu złe.

To informuję pana marszałka, że Wysoki Sejm jest w czerwonej strefie i ludzie, którzy dzisiaj oglądają nasze obrady, robią to nielegalnie. Takie są przepisy, które wprowadzacie. To jest rozporządzenie z piątku.

Znaleźliśmy też bezpodstawne rozróżnienie lekarzy na lepszych i gorszych. Okazuje się, że ta ustawa wyeliminowała 70% medyków, jeśli chodzi o dodatki do ich pensji. Ta ustawa nie zajęła się też personelem medycznym. Ludzie, którzy pracują w szpitalach na oddziałach zakaźnych, którzy obsługują sprzęt, w tej ustawie po prostu zostali pominięci. Właśnie z tego powodu: żeby opinia publiczna nie dowiedziała się, jak wiele w tej ustawie jest błędów i jak wiele osób w tej ustawie zostało po prostu pominiętych. Tu też będzie nasza poprawka. Chcecie, żeby zamiast dyrektorów szpitalami zarządzali partyjni nominaci w stylu Jacka Sasina. Nie będzie na to naszej zgody, absolutnie nie.

To są projekty przygotowane, które powinny być wprowadzone dawno temu, bo one leżą w Wysokiej Izbie od dłuższego czasu. Wysoka Izbo! Nauka płynie z tego prosta: nad prawem warto pracować dłużej niż kilka godzin. To jest wasza dziesiąta ustawa w sprawie COVID-u. Sami w tej ustawie zmieniacie przepisy, które zmienialiście jeszcze chwilę temu. 2–3 miesiące temu np. wprowadzaliście odpowiedzialność lekarzy, chcieliście ich karać za błędy, których nie popełnili specjalnie. Dzisiaj od tego odchodzicie. Przecież państwo za tym głosowali. To wy wprowadzaliście te zmiany. To po co robić kolejną ustawę na kolanie, jak można nad tym spokojnie pracować?

Wysoka Izbo! Prawda jest taka, że ten rząd po prostu bierze pełną odpowiedzialność za sytuację w Polsce. Nie wiem, czy jest z nami pan minister Kraska, wiceminister zdrowia, jeden z waszych głównych specjalistów do spraw COVID-u. Pan minister Kraska 6 tygodni temu: Druga fala koronawirusa będzie łagodniejsza.

Jeżeli ktoś dzisiaj mówi o szpitalach na stadionach, to wynika to właśnie z takich opinii. Minister Dworczyk wczoraj: Druga fala koronawirusa jest dużo większa. No jest dużo większa, faktycznie, niż mówili wasi eksperci, i dlatego jesteśmy do tego nieprzygotowani jako państwo. Trzeci cytat, pan premier Morawiecki: Zwalczyliśmy tę chorobę. Jesteśmy liderami w Europie. Jesteśmy liderami w Europie, to prawda. Tylko zastanawiam się, co pan premier robił wczoraj na konferencji na tle respiratorów, bo moim zdaniem uprawiał tam po prostu propagandę. Gdzie był pan premier w ciągu 6 miesięcy, kiedy te respiratory były tak potrzebne? Nowa ustawa, o której mówimy dzisiaj - to jest właśnie złudne myślenie, że w momencie kryzysu wystarczy napisać na papierze, że będzie dobrze. Właśnie tam są takie zapisy, że szpital musi przyjąć, że karetka musi zawieźć. Ale przecież do tej pory na papierze też się wszystko zgadzało, przecież była wystarczająca liczba łóżek, wystarczająca liczba respiratorów, a na samym końcu okazało się, że jednak tak nie jest, że karetki odbijały się od szpitali, bo zmarnowaliście 6 miesięcy. Ktoś wczoraj mądrze to określił, że zamiast walką o łóżka zajmowaliście się walką o stołki. I taka jest prawda, jeżeli chodzi o ostatnie 6 miesięcy. Samorządy. Dzisiaj samorządy biorą na siebie ciężar. Pytanie do wnioskodawcy, pana posła Protasa: jak wielkie jest zaangażowanie samorządów, które odciąża dzisiaj rząd? Tam nie ma odpowiedzi na te pytania, tam nie ma rozwiązań. W związku z tym chciałbym też zapytać. Mówicie, że ściągniecie lekarzy z zagranicy, tych lekarzy, o których pani poseł Hrynkiewicz z tej mównicy mówiła: „niech jadą” Tych lekarzy chcecie ściągnąć z zagranicy? Ci lekarze już dawno tam są. Oni dzisiaj wyjechali. Dzisiaj chcecie ich ściągać, dzisiaj się obudziliście? Nie ma go tu dzisiaj, ale mam nadzieję, że nas słucha, mimo że to nielegalne.

Albo rodzinie pana Tadeusza z Mirostowic? 68 lat, przez tydzień był leczony na przeziębienie. Okazuje się, że miał COVID, nie trafił pod respirator i zmarł. I wreszcie taka historia, która każdego z nas bardzo mocno uderzyła: Bartek, lat 17, źle się czuł, zapadł w śpiączkę, lekarze podejrzewali koronawirusa, więc jeden szpital go nie przyjął, odesłali go do innego, gdzie czekał 10 godzin na przyjęcie. Nie miał koronawirusa, miał ropień śródczaszkowy. Zmarł 2 dni po operacji. I nie chcemy dzisiaj słyszeć od was fałszywych zapewnień. Nie chcemy słyszeć tych tekstów pana ministra Szumowskiego, który mówił, że jesteśmy przygotowani na każdy wariant i on teraz może jechać na wakacje. Chcemy, żeby Polacy mogli usłyszeć, jaka jest prawda o tej chorobie i o epidemii, jaki jest stan epidemii, co nas czeka w najbliższych tygodniach. I że wszystko jest pod kontrolą, budują się nowe stadiony, hale, szpitale. Przez pół roku kłamaliście i chcemy wiedzieć, jakie są oficjalne prognozy, ile osób może być chorych, ile osób może umrzeć, dla ilu osób może zabraknąć miejsc w szpitalach, ile zabraknie respiratorów. To są pytania, na które musicie odpowiedzieć opinii publicznej. Jaka jest strategia walki z COVID-em? Ile może być zachorowań w ciągu najbliższych tygodni? Jesteście jedynym rządem w Europie, który ukrywa te dane przed obywatelami. My tego nie wiemy, nie wiemy, jak wirus się będzie rozwijał, bo nikogo o tym nie informujecie, mimo że macie wszelkie możliwe służby i że możecie ich użyć. Nie wiemy, co będziecie robili ze szkołami, nie wiemy, co będziecie robili z restrykcjami. Po prostu powiedzcie prawdę, bo nie jesteśmy w TVP Info. Tu nie wystarczy pudrowanie rzeczywistości. Potrzebna jest rzetelna informacja dla wszystkich. Przez ostatnie 5 lat w jednym byliście bardzo sprawni, w zdobywaniu dla siebie władzy. Nic wam tak dobrze nie wyszło. Zaczynaliście tutaj, w parlamencie, później były trybunały, sądy, spółki, media. Wymieniliście dziesiątki tysięcy wspaniałych urzędników na nominatów partyjnych. Zatrudniliście swoich synów, swoje córki, swoich wujków, sąsiadów, wszystkich zatrudniliście. I macie całą tę władzę, o której marzyliście - całą tę władzę. Przez ten jeden moment. Zdobyliście ją całą. Polacy dzisiaj liczą na to, że wykorzystacie tę władzę w dobrym celu. Jak ją wykorzystaliście w ciągu tych 6 miesięcy? Widzę tylko, że zmarnowaliście po prostu czas, czas nas wszystkich, czas milionów Polaków, którzy dzisiaj czekają na solidne rozwiązania. Państwo, które stworzyliście, jest po prostu chore, to jest państwo PiS. Jak w soczewce widać dzisiaj wszelkie możliwe problemy. To państwo musi być zdrowe, bo to jest nasze państwo. I każdy Polak, i każda Polka musi wiedzieć, że może liczyć na swój rząd. I ostatnie zdanie, panie marszałku, jeśli pan pozwoli. Pan premier Morawiecki zwracał się wczoraj z apelem do Senatu, [[Dzwonek]] żeby nad tą ustawą procedowano szybko. Jeżeli my nad tą ustawą będziemy procedować dobrze w Sejmie, jeżeli poprawki Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy zostaną przyjęte, to nie będzie konieczności, żeby nad tą ustawą pracować w Senacie. A więc ja apeluję do większości sejmowej: pracujmy nad tą ustawą, przyjmijcie dobre poprawki ten jeden, jedyny raz, bo one są po prostu potrzebne, i zamknijmy tę sprawę jak najszybciej, żeby ta ustawa była po prostu dobra, a nie byle jaka. Muszę to powiedzieć, że to dzięki panu opóźniliśmy prace o 1 dzień. Tylko polityczne ględzenie.

Już skończyliście państwo przerzucać się oskarżeniami? Świetnie. Wysoka Izbo! Otóż, panie premierze, panie ministrze zdrowia, strategii na jesień nie ogłasza się jesienią, tylko na początku lata. Strategia to nie tylko plan na miesiąc czy dwa, ale wszystkie scenariusze, te dobre i te złe. Strategii wreszcie nie zmienia się co 2 tygodnie, tak samo zresztą jak czterech ustaw nie przekazuje się posłom na 17 godzin przed ich zbiorczym procedowaniem w Sejmie. Projekty te powinny być konsultowane ze środowiskiem medycznym i ekspertami, opozycja powinna mieć czas na rzetelne przygotowanie poprawek i ich konsultację. My naprawdę widzimy wasze trudności i chcemy wam pomóc. To dotyczy nas wszystkich, wszystkich obywateli. Jedną z kluczowych kwestii od początku pandemii, czyli, lekko licząc, od 6 miesięcy, jest opanowanie liczby zakażeń i wygaszanie ognisk choroby. Sanepid alarmował już wiosną, że nie wyrabia się z pracą. Obecnie odbiera tysiące telefonów. Ludzie narzekali, że nie mogą się dodzwonić do sanepidu przez wiele dni. Przez pół roku nie zrobiliście z tym nic. Proponujecie zatrudnienie większej liczby zastępców głównego inspektora sanitarnego - musztarda po obiedzie. Lewica nie będzie sprzeciwiać się temu rozwiązaniu, ale sanepid potrzebuje dziś przede wszystkim rąk do pracy, ludzi do odbierania telefonów, udzielania informacji, śledzenia kontaktów osób zakażonych, a nie tylko kilku dodatkowych dyrektorów. Dlatego już tydzień temu na spotkaniu z rządem wśród wielu innych propozycji my proponowaliśmy zaangażowanie do realizacji tych zadań firm prywatnych. Wszystkie narzędzia macie w ręku. Nie potrzeba na to dodatkowych środków, nie potrzeba na to dużo więcej czasu. Wszystkie narzędzia macie w ręku. Po prostu to zróbcie. Według naszych szacunków da nam to od 5 do 20 tys. nowych stanowisk konsultacyjnych, które mogą wesprzeć nas w walce, w zakresie ograniczania choroby. Złożyliśmy tu ustawę, która nareszcie daję podstawę prawną do nakazu noszenia maseczek przez wszystkich obywateli. Da ona organom państwa niezbędne uprawnienia, których zabrakło w poprzednich tarczach antykryzysowych, ale pozwoli też bronić pracowników firm usługowych czy sklepów, którzy wreszcie będą mogli odmówić obsługiwania klientów, którzy maseczek nie noszą. Liczymy na jej poparcie przez koalicję rządzącą i opozycję. Przez ostatnie 6 miesięcy, kiedy radośnie wprowadzaliście i likwidowaliście szpitale jednoimienne, dawaliście i zabieraliście dodatki za pracę w związku z COVID, a pan premier obwieszczał koniec pandemii, liczba zakażeń systematycznie rosła, potem rosła gwałtownie, a dziś szybuje w górę w zastraszającym tempie. Dziś, gdy system opieki medycznej właściwie już się załamał, a szpitale przepełnione i pozbawione lekarzy odsyłają pacjentów, wy zaczynacie dopiero organizować dodatkowe ręce do pracy. I znowu chce się rzec: musztarda po obiedzie. Lewica oczywiście jest za częścią rozwiązań, które znajdziemy w ustawie, którą tu dzisiaj omawiamy, za tym, aby wszystkim pracownikom opieki medycznej za okres kwarantanny przysługiwało 100% wynagrodzenia, ale muszą one objąć wszystkich pracowników, niezależnie od rodzaju umowy, także tych pracujących na kontrakcie czy zatrudnionych przez firmy zewnętrzne, także salowe i laborantów.

Jesteśmy za podniesieniem kwot za skierowanie do pracy w związku z pandemią do 200%, ale te dodatki powinny przysługiwać także tym pracownikom ochrony zdrowia, którzy już z pandemią walczą, nie tylko tym, którzy zostaną do tej walki skierowani. I tu też złożymy odpowiednią poprawkę.

Postulujemy odejście od kar bezwzględnego więzienia za błędy medyczne. Dziś jest dzień, w którym trzeba cofnąć zmianę art. 37a Kodeksu karnego, bo czas przestać karać lekarzy, czas przestać ich obwiniać za wszystko, a trzeba ich zacząć wspierać. I odpowiednią poprawkę również dziś złożymy. Ostatnie 6 miesięcy to był czas na regulacje dotyczące budowy szpitali polowych, ustaleń zasad pracy lekarzy, szkolenia personelu i mobilizowania dodatkowych sił do pracy. Był czas na konsultacje ze środowiskiem medycznym, był czas na szkolenie i mobilizowanie studentów i przedstawicieli innych zawodów medycznych i okołomedycznych. Proponujecie te rozwiązania dopiero dziś - musztarda po obiedzie. Przepisy dotyczące powoływania lekarzy są niedopracowane i wewnętrznie sprzeczne. Pozwalają na powołanie rodziców najmłodszych dzieci, a nawet matek karmiących. Lewica nie zagłosuje za takimi rozwiązaniami i również złoży odpowiednie poprawki. Twierdzicie, że idziemy drogą środka, że są jeszcze dostępne łóżka i respiratory, choć szpitale jasno mówią co innego i fizycznie nie mają gdzie przyjmować pacjentów. Chcecie powoływać koordynatorów - musztarda po obiedzie. Czas na koordynację był pół roku temu, a nie teraz. Teraz nie ma czasu na uciekanie od odpowiedzialności. i zrzucanie decyzji na szpitale i ratowników. Pozostawiliście ich samym sobie. Dziś na łapu-capu wprowadzacie stanowisko superkoordynatora ratownictwa medycznego, który kolanem będzie upychał pacjentów, gdzie się da. Koordynator nie wyczaruje miejsc w szpitalach, nie stworzy z powietrza respiratorów, nie wyczaruje nowych lekarzy i pielęgniarek. A za odmowę wykonania polecenia grozicie szpitalowi odwołaniem dyrektora, co w warunkach epidemii i spowodowanego nią przeciążenia wywoła tylko jeszcze większy chaos. Jesteśmy natomiast za prawem pacjentów do równego traktowania. Lepiej późno niż wcale. Mam nadzieję, że ból posłów Czarnków, Szumowskich i Kaczyńskich nie będzie już nigdy większy niż ból zwykłych obywateli. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewicy. Wysoka Izbo! Mamy wypracowane już mechanizmy, procedury, szpitale jednoimienne, gotową sieć laboratoriów, testy genetyczne, szybkie testy na czas jesienny, by zdiagnozować możliwe zakażenia - to wszystko jest przygotowane. Przygotowałem rekomendacje na jesień, które są bardzo proste, spójne, możliwe do wdrożenia. Przygotowałem wszystkie plany na jesień. Myślę, że mój następca będzie je wdrażał w sposób bezpośredni. Myślę, że pan poseł Szumowski nas ogląda. Otóż, panie pośle, minister Niedzielski chyba zgubił kluczyk do biurka, w którym pan zostawił te wszystkie rekomendacje, i po prostu tego nie wdrażał. Wczoraj w telewizji publicznej czytaliśmy: opozycja blokuje walkę z pandemią, opozycja gra życiem i zdrowiem Polaków. Nie będę komentował tych głupstw, ale muszę skomentować słowa pana ministra zdrowia, który w ramach partyjnego przekazu twierdził we wszystkich mediach, że jego wczorajszą absencję tutaj, w Wysokiej Izbie.

Otóż, panie ministrze, nie. Niech pan, cytując klasyka, nie idzie tą drogą. My daliśmy panu czas, by zapoznał się pan z uwagami do ustawy, które przedstawiły Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. I mam propozycję do pana, panie ministrze zdrowia. Niech pan dzisiaj tutaj, w Wysokiej Izbie, przedstawi stanowisko odnośnie do tych ważnych uwag, które przedstawiły te podmioty. Pracownicy i pacjenci służby zdrowia zarzucają projektowi ministerstwa obniżenie standardów i niewykonalność. Niewykonalność to nakazanie samorządom zawodów medycznych, aby w ciągu dnia, 7 dni przekazały wykaz osób, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Być może pan minister jeszcze tego nie wie albo nie czytał tej swojej ustawy o dobrym samarytaninie, jak to określa, ale samorządy zawodów medycznych gromadzą tylko te dane osobowe i wrażliwe, które są określone właściwymi ustawami. Chciałem pana zapytać: Czy jeden dzień zwłoki w Sejmie tak ogromnie spowalnia prace?

Boję się tego, dlatego że w ramach tej kluczowej roli inspekcji mamy zwiększenie o dwie osoby kierownictwa Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Przypomnę też, że jeszcze miesiąc temu informował nas on, że wszystko to ulega wypłaszczeniu. Wtedy kiedy Polacy już walczyli z epidemią, to sanepid walczył o to, jak zlikwidować u siebie strukturę, która była strukturą sanepidowską, w służbach wewnętrznych, w Policji i w Służbie Więziennej. Dzisiaj pracownicy sanepidów są przemęczeni [[Dzwonek]] fizycznie i psychicznie. I pytają: Czy pan premier wzmocni tę służbę o pracowników, którzy tracą pracę w administracji rządowej?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Najpierw dobre słowo do wszystkich, którzy walczą z epidemią, do wszystkich pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarek, ratowników. Wiemy, w jakich pracują warunkach. Te cztery projekty poselskie - bo nie tylko ten jeden, o dobrym samarytaninie, został złożony do Wysokiej Izby - są przedmiotem dzisiejszych obrad. W tym również klub Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 złożył projekt mówiący o tzw. premii dla bohatera, o wynagrodzeniu pracowników służb zdrowia, którzy pracują na rzecz tych, którzy potrzebują pomocy. Projekty te są ważne, zgadzam się tutaj z panem ministrem zdrowia, natomiast nie mogę się zgodzić z jego oceną, że politykierstwo wygrało ze zdrowiem. Rozumiem, że pan minister jest przywiązany do swojego projektu, bo de facto ten projekt poselski jest projektem rządowym, i mówi, że te projekty nie budzą kontrowersji. No to ten wczorajszy dzień pozwolił nam na zapoznanie się ze stanowiskiem Naczelnej Izby lekarskiej, która jest zaniepokojona i rozczarowana projektem. Cytuję: spodziewaliśmy się wsparcia, a w regulacjach znajdujemy odbicie nieprzyjaznych wypowiedzi polityków.

Samorządy. Wskazanie czterooddziałowego szpitala powiatowego jako miejsca, gdzie ma być prowadzona walka z COVID-em, gdzie mają być leczeni ci pacjenci, to de facto wygaszenie prawie wszystkich jego oddziałów.

Wydaje mi się, że. Jak samorząd ma później zarządzać szpitalem, który poniesie ewentualne straty finansowe?

Ustawa jest w jego opinii przygotowana z dnia na dzień, a było tyle czasu. Mówi też, że decyzje rządu związane z epidemią potężnie zachwiały zaufaniem społecznym. To mówi przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy.

Przynajmniej literalnie z tego przepisu to nie wynika. Przecież analizowali go również przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej i związków zawodowych.

Trzeba mieć rezerwy, tylko można było to zrobić wcześniej.

Może to zwiększyć dostępność usług medycznych, ale trzeba włączyć finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Złożymy odpowiednie poprawki.

Przecież to jest niezmiernie ważna kwestia. Premia dla bohatera, dobrowolny ZUS i przede wszystkim zregionalizowane podejście do zwalczania epidemii.

Kontynuuje pan poseł Jarosław Rzepa. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Wiele samorządów wojewódzkich ma w swoim obszarze funkcjonowania uzdrowiska, które mają odpowiednią bazę, w których pracują ludzie: lekarze, pielęgniarki.

Bardzo dziękuję wszystkim za propozycje, choć w wielu przypadkach wydaje mi się, że szkoda, że rządzący nie wysłuchali ich wtedy, kiedy był na to czas.

Nie, szanowni państwo. Dzisiaj trzeba zapłacić tym ludziom, którzy robią to od wielu miesięcy. Zadbaliście państwo w tym projekcie ustawy o Policję, Straż Graniczną, SOP. Dobrze, że nie zapomnieliście o medykach, ale gdzie są ci ludzie, którzy od samego początku to robili?

Jeżeli w jakikolwiek sposób nie przyjmą.

Szanowni Państwo! Kto odpowie za błędy państwa pełnomocników? Dodatkowo jeszcze uchylacie choćby rady społeczne tych szpitali. One nie będą miały nic do powiedzenia. Szanowni Państwo! Mam nadzieję, że przyjmiecie państwo te poprawki. Dzisiaj na posiedzeniu Komisji Zdrowia wprowadzimy szereg poprawek i chcemy wspólnie zrobić to, o czym mówimy. Są merytoryczne, pani poseł. Wysłuchacie przede wszystkim w imieniu ludzi, którzy dzisiaj obserwują, którzy mówią, że nie chodzi tylko o to, żebyście państwo wymagali od nich listy w ciągu 7 dni.

Nie prowadzą, szanowni państwo. Szanowni Państwo! My jako klub Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego deklarujemy, że chcemy współpracować, ale na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Zdrowia powiemy: wielkie sprawdzam.

Jeden z moich przedmówców powiedział: panie premierze, trzeba myśleć do przodu. Do przodu, i to daleko. Niestety mam w wielu przypadkach świadomość, że te działania są tylko i wyłącznie o krok przed nami. Dziękuję serdecznie. Witam państwa z wielką przyjemnością. Zapraszam pana posła Dobromira Sośnierza z Koła Poselskiego Konfederacja. Panie pośle, mównica jest pana. Nie daję jej panu, tylko zapraszam. I mam prośbę, żeby pani nie komentowała, bo zaraz wezwę marszałek Witek i będzie pani zastrachana. Proszę bardzo, panie pośle. Wiemy już, że jesteśmy w czarnej... dziurze, gorzej, że najwyraźniej zaczynamy się w niej pomału urządzać. To jest kolejna specustawa COVID-owa, która świadczy o tym, że rząd zamiast szybko z tej dziury wyłazić, rozstawia w niej pomału meble. Wszystkie te regulacje pokazują, że epidemia zaplanowana jest według rządu na dłużej i dlatego w tej doraźnej partaninie ustawodawczej kilka trytytek musimy teraz wymienić na grubsze, musi to jeszcze trochę postać. Projekt zapowiada na przykład zniesienie odpowiedzialności lekarzy na czas epidemii, a dopiero co w jednej ze słynnych tarcz zaostrzaliśmy tę odpowiedzialność. Czyżbyśmy znowu wyrypali się o własne nogi?

A teraz zamiast wycofać się z tego niepotrzebnego przepisu, produkujecie kolejny, który będzie doraźnie usuwał jego skutki, z dużymi znamionami przedobrzenia w drugą stronę.

Wmontowujecie w cały system wadliwe mechanizmy, które zachęcają do naciągania statystyki produkowania różnych fałszywych przypadków i dlatego np. rodzice nastolatka z rozciętą twarzą są zmuszani do podpisania oświadczenia, że podejrzewają u niego COVID.

Za pieniądze wydane na miliony mało wiarygodnych testów moglibyśmy, nie wiem, postawić kilka szpitali albo zatrudniać personel. Wiele innych chorób zakaźnych leczymy bez masowych testów, i to całkiem skutecznie, więc po co to robicie. Muszę zostawić czas kolejnemu mówcy, przepraszam. Zapraszam pana posła Michała Urbaniaka.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Otóż żywię nadzieję, że dostatecznie Izba przemyślała sprawę tych nowiutkich multiustaw, które są przygotowywane. Odniosę się głównie do Prawa i Sprawiedliwości - proponujecie państwo nieprzemyślane rozwiązania, a jeśli już znajdzie się coś sensownego, to zdecydowanie za późno i oczywiście w ramach akcji wielosztuków po raz kolejny. Idea jest oczywiście słuszna, ale nie dziwię się, że proponują państwo taki zapis, ponieważ zaniedbaliście przez ostatnie lata bezpieczeństwo lekowe, produkcję leków w Polsce. Leki w większości ściągane są z Azji. Dlaczego nie wspieraliście produkcji leków i substancji aktywnych w Polsce? W końcu mamy sytuację, w której pracownicy służby zdrowia czy pracownicy mundurowi dostaną 100% zasiłku chorobowego w sytuacji, w której ci państwo będą pracować z COVID, zostaną zarażeni bądź pójdą na kwarantannę. Słusznie, szkoda, że dopiero teraz, a nie kilka miesięcy temu, o czym mówiliśmy już dawno. Mówią państwo o środkach ochrony osobistej, ale sami nie zwiększacie ilości tych środków dla medyków. Nie macie przygotowanych miejsc noclegowych dla medyków w sytuacji, w której ktoś zostałby zarażony, a nie chciałby narażać także swojej rodziny. Mówicie o zapisie o dobrym samarytaninie. Problem w tym, że rozszerzając ten zapis, wprowadziliście chaos prawny, a dużo lepiej byłoby rozszerzyć tylko taki zapis np. dla studentów, którzy idą pracować przy COVID-zie. W ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty ponownie chcecie wprowadzić zapis o dopuszczeniu cudzoziemców do wykonywania zawodu lekarza bez nostryfikacji dyplomu. Po raz kolejny próbujecie wprowadzić tylnymi drzwiami zapis, który mówi jasno o tym, że nie jesteście [[Dzwonek]] przygotowani na COVID-19 ani na żadne inne choroby. Bo jeśli dzisiaj będziemy ściągać, przykładowo, jakichś lekarzy bądź medyków, bądź pielęgniarki chociażby ze Wschodu, to jaką mamy gwarancję, że te dyplomy nie były kupione na targu? Żadnej. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, przechodzimy do zadawania pytań. Przypominam, że tych pytań łącznie jest 30. Każdy klub wie, ile może zadać pytań.

Damy radę. Wysoka Izbo! W dniu wczorajszym posłowie opozycji w mediach ogólnopolskich, z ogólną determinacją chcąc zdyskredytować przedłożenie z druku nr 683, udzielali informacji na antenach naprawdę o dużej oglądalności, iż są w tej ustawie zapisy, które spowodują, zacytuję, że kobieta, która urodzi dziecko - lekarz, pielęgniarka - po 2 dniach może być skierowana do pracy. To jest naprawdę draństwo, co państwo robicie, to jest uderzenie w podstawowe. Bardzo proszę, żeby przedstawiciel wnioskodawców tego druku sejmowego wytłumaczył Wysokiej Izbie, jakie są zapisy w art. 14 ust. 4, i zdementował tę potworną. Dziękuję serdecznie. Zapraszam panią poseł Monikę Wielichowską z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzięki temu, że wczoraj do pracy nie przyszli Kaczyński, Morawiecki, Ziobro, Gowin i 24 innych posłów Zjednoczonej Prawicy, mieliśmy czas na dobrą legislację. To ważne, bo [[Oklaski]] każdy projekt ustawy powinien wpisywać się w jasną i spójną strategię rządu dotyczącą walki z pandemią, strategię, która powinna być przemyślana, konsekwentna, komunikowana i realizowana. I musi być ona dobrze przygotowana, ale, choć musi, nie jest, bo wszystkie projekty piszecie, drodzy państwo, na kolanie, ekspresem przepychacie w Sejmie bez konsultacji społecznych. Chaos w służbie zdrowia jest coraz większy, strach obywateli pogłębia się każdego dnia i wszystkich nas dotkną, wszystkich nas, surowe tego konsekwencje. Dlatego tak ważne jest, by już zaprzestać procedowania (Dzwonek) złych ustaw, złego prawa, ponieważ najważniejsze jest zdrowie, życie i bezpieczeństwo obywateli. Ja bardzo ubolewam, że dzisiaj na sali nie ma pana ministra Niedzielskiego, który nie znalazł czasu na dzisiejszą dyskusję, debatę, ale znalazł czas wczoraj, żeby wypisywać bzdury w mediach społecznościowych, choć powinien nam, opozycji, podziękować. Za co? ...za to, że chcemy tworzyć dobre prawo. Bo nie czarujmy się, to jest ustawa rządowa, która jest oczywiście przepychana poselskim schematem, żeby uniknąć konsultacji społecznych i dobrego procedowania, jak powiedziałam na wstępie. Dziękuję bardzo. Będziemy się łączyli z panią posłanką Marceliną Zawiszą, która zdalnie będzie zadawała pytania. Witamy panią posłankę. Wysoka Izbo! Jak rząd zamierza poradzić sobie z leczeniem pacjentów z innymi niż COVID chorobami? Przekształcenie miejsc szpitalnych i budowa szpitali polowych będzie pochłaniała przecież zasoby. Już mamy zaległości choćby z przesuwanymi zabiegami planowanymi, pacjenci po transplantacji zgłaszają problemy z dostępem do ochrony zdrowia, diagnostyka raka piersi czy raka szyjki macicy leży. Ta ustawa nie daje odpowiedzi na te palące problemy, proszę więc rząd o odpowiedź na pytanie, jak zamierzacie sobie z tym poradzić. Nie ma w tej ustawie też jasnego rozwiązania kwestii wynagrodzeń dla osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii, pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Czy dodatkowe wynagrodzenie przysługujące w tych wypadkach będzie liczone względem realnych dochodów tych osób? Dlaczego podwyżka nie obejmuje pracowników sanepidu, którzy pracują ponad swoje siły?

Zapraszam pana posła Dariusza Klimczaka z Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Chciałbym zapytać o zmiany w systemie ratownictwa medycznego. Mianowicie próbujecie wzmocnić rolę koordynatora wojewódzkiego, powołujecie, tworzycie nową funkcję koordynatora krajowego. Czy żeby znaleźć wolne łóżko w naszym kraju, trzeba powoływać nowy urząd? Przecież każdy szpital ma system, w którym widać, czy łóżka są wolne, czy zajęte. Co za problem, żeby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia skoordynowało to i żeby ten system służył do znajdowania wolnych łóżek? Trzeba powoływać nowy urząd? Co wy chcecie ukryć, próbując w ten sposób, ręcznie, na siłę sterować wolnymi łóżkami? Druga sprawa. Przecież każdy z nas korzysta z Internetu. Kiedy kupuję dany produkt, osoba na drugim końcu kraju wie, że tego produktu nie ma. Przecież to jest abstrakcja. Następnie teleporady. Kiedy wreszcie skończycie z tym systemem, w którym ludzie (Dzwonek) odbijają się od lekarza? Przecież teleporada powinna być dostępna dla człowieka, który kontynuuje leczenie. Ten, kto ma nową dolegliwość, powinien mieć dostęp do lekarza. Telekontrole wprowadźcie sobie w skarbówce albo w innych urzędach, żeby nie dotyczyły przedsiębiorców, ale w sprawie zdrowia pacjent powinien mieć dostęp do lekarza. Zapraszam pana posła Artura Dziambora z Koła Poselskiego Konfederacja. Mam dwie sprawy. Nad tym dzisiaj będziemy procedować i prawdopodobnie koalicja Lewicy z Platformą i PiS-em wprowadzi zakaz, a właściwie nakaz noszenia maseczek.

Moje pytanie brzmi: Czy zostaną one anulowane? To jest o tyle ważne, że ze strony władzy byłby to gest uczciwości wobec tych wszystkich obywateli, którzy po prostu przestrzegali prawa (Dzwonek), którzy byli zmuszani do tego, żeby nosić maseczki, przez policję, pod groźbą kary, a ta kara była nielegalna.

Jeżeli ten projekt wejdzie w życie bez poprawek, może się okazać, że przedsiębiorca, który np. nie założył maseczki, będzie pozbawiony pieniędzy z tarczy i ucierpią wszyscy jego pracownicy. Takie absurdy on zawiera.

W imieniu Polski 2050 złożę poprawki i bardzo proszę o ich przyjęcie. Dziękuję bardzo.

Szanowni państwo, naprawdę w tej sprawie musimy działać wspólnie. Część tych złośliwych, niepotrzebnych głosów, które padały, niczego pozytywnego nie wnosi, tym bardziej że też macie państwo w swoich projektach dobre rozwiązania, które są również w projekcie Prawa i Sprawiedliwości, a więc pracujmy razem. A pana ministra chciałem zapytać o te nieprawdy, które były powtarzane wczoraj w mediach, które były mówione z tej mównicy. Warto też powiedzieć chociaż dwa zdania o zwiększeniu finansowania pracowników, o [[Dzwonek]] klauzuli dobrego samarytanina i innych dobrych rozwiązaniach. Dziękuję serdecznie. Teraz z ciekawością wysłuchamy pytania zadanego przez panią posłankę Barbarę Nowacką z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Spróbuję sprostać, aczkolwiek właściwie puste ławy rządowe i kilku etatowych krzykaczy ze strony PiS-u pokazują szacunek dla tematu. A państwo najpierw przygotowujecie bubel, a potem nawet nie chcecie przyjść i o tym podyskutować. Mówicie o sobie: Prawo i Sprawiedliwość. No to gdzie prawo rodzin do zajęcia się malutkim dzieckiem, które w waszej ustawie zostało wykasowane? Gdzie sprawiedliwość dla medyków, którzy są różnicowani pod względem wynagrodzenia? Zapominacie o ratownikach medycznych, salowych, o wszystkich, którzy pracują w ochronie zdrowia. Każdy z nich będzie się stykał z COVID-em, każdy z nich jest narażony, oni i ich rodziny, a wy mówicie wyłącznie o tych kierowanych przez wojewodę. Wywołujecie wojny w środowisku medycznym, zamiast realnie pomóc. Wynagrodzenia [[Dzwonek]] powinny trafić do wszystkich, równo i sprawiedliwie, do wszystkich, którzy walczą na froncie zdrowia. Wy polegliście, wy zawiedliście. Te wasze prawo i sprawiedliwość okazały się fałszem. Zapraszam panią posłankę Monikę Falej, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Karetki z pacjentami, także tymi wymagającymi natychmiastowej pomocy, jeżdżą od szpitala do szpitala. Lekarze coraz rzadziej zajmują się pacjentami, bo większość czasu spędzają przy telefonie, szukając wolnych miejsc w szpitalach. Rząd wysyła lekarzom, pielęgniarkom nakazy pracy, nie robiąc nic, aby wprowadzić system, który będzie gromadził takie dane i informacje. W projekcie ustawy przewidziano podwyżki dla lekarzy, i to jest dobry krok, co prawda spóźniony o wiele miesięcy, ale mimo wszystko dobry. System ochrony zdrowia to jednak nie tylko lekarze, ale także pracownicy i pracownice medycznych laboratoriów diagnostycznych. Przywykliśmy już do tego, że dzielicie ludzi na sorty, ale do tej pory kryterium były poglądy, a teraz do gorszego sortu zaliczyliście diagnostów laboratoryjnych i techników analitycznych [[Dzwonek]] analityki medycznej. W czym oni wam zawinili? Dziękuję serdecznie. Wysoki Sejmie! Przykre to, że nawet w sytuacji epidemii, kiedy wszyscy powinniśmy działać razem, opozycja nie potrafi odstąpić od politycznej walki. Pokazaliście państwo wczoraj, że nie potraficie działać w sytuacji podwyższonej konieczności, w sytuacji pilności podejmowania działań i sypiecie piasek w tryby nawet wtedy, kiedy konsekwencje waszych działań uderzają w Polaków. Mówiliście, że nie znacie ustawy, ale nie przeszkadzało to wam nazywać ją kamaszową, mimo że podobno nie znaliście jej treści. Tymczasem jest to ustawa dobrego samarytanina, wspierająca medyków i wzmacniająca działania w walce z epidemią. Posłowie opozycji manipulują, nawet teraz, kiedy podobno przeczytali tę ustawę, manipulują, szerzą fake newsy i Mam pytanie do pana posła przedstawiciela wnioskodawców. Panie pośle, jakie regulacje wspierające medyków w walce z epidemią zawarte są w tej ustawie i dlaczego trzeba ją uchwalić? Mam prośbę do opozycji: Wyjdźcie wreszcie z politycznej piaskownicy. Nie czas na polityczne walki, tylko czas na wspólne działanie dla zdrowia i bezpieczeństwa Polaków. Teraz pytanie zada pan poseł Robert Kropiwnicki z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Otóż zarzuca nam się, że politykujemy. My dbamy o zdrowie Polaków, bo wy dawno o tym zapomnieliście.

To jest skala waszych zaniedbań. Mieliście na to 8 miesięcy i roztrwoniliście ten czas, bo walczyliście o to, kto będzie ministrem, kto będzie prezesem spółki, gdzie zatrudnicie swoje dzieci. To było dla was ważniejsze niż ratowanie zdrowia i życia Polaków. Pytam: Co zrobicie, jak pomożecie pracownikom sanepidów, jak pomożecie ratownikom medycznym? System ochrony zdrowia rozsypuje się na naszych oczach, a wy radośnie mówicie, że będziecie budować nowe szpitale. Pomóżcie tym, którzy są już dzisiaj, pomóżcie ratownikom medycznym, pomóżcie pogotowiom ratunkowym, bo oni dzisiaj naprawdę cierpią, a oni są na pierwszej linii frontu. Ta ustawa to jest jeden wielki bubel. Oczekiwaliśmy wielkiej strategii, bo był czas na to, żeby ją przygotować, a wy przynieśliście bubel, który się do niczego nie nadaje. Kupa kamieni przy tym, co wy przynieśliście, to jest wielka konstrukcja budowlana. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana posła Dariusza Wieczorka z klubu parlamentarnego Lewicy. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście dzisiaj dyskutujemy nad czterema projektami ustaw i pewnie skończy się to tak, że ostatecznie po południu będziemy mieli do czynienia z jednym projektem ustawy. Mam nadzieję, że zapisy, które są w tych pozostałych projektach przygotowanych przez opozycję, w tym jednym projekcie również się znajdą. Prawda jest taka, że w tym projekcie mówimy o środkach finansowych, które będą przekazywane na rzecz tych, którzy będą kierowani przez wojewodów do w pracy w zwalczaniu epidemii. Natomiast rzeczywiście jest bardzo poważny problem dotyczący pracowników pogotowia ratunkowego, dotyczący laborantów, dotyczący wszystkich tych, którzy funkcjonują dzisiaj w ochronie zdrowia. Pytanie do projektodawców jest takie: Czy macie w tym zakresie przeprowadzone analizy i czy przewidujecie, jeżeli chodzi (Dzwonek) również o pozostałych pracowników ochrony zdrowia, rekompensatę i podwyżki? Zapraszam panią posłankę Agnieszkę Pomaską z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie i Panowie Posłowie! Minister Niedzielski dziwi się, że niektórzy szukają pomysłu, jak obejść obostrzenia. Panie ministrze, ludzie szukają pomysłu, jak obejść obostrzenia, bo wam już po prostu nie ufają, ludzie nie ufają tej władzy. Bo jak mają ufać tej władzy, wtedy kiedy premier Morawiecki mówi, czego nie można w restauracjach, a sam te zakazy łamie? Wtedy kiedy premier Kaczyński pojawia się publicznie bez maseczki, wtedy kiedy kupowane są respiratory od handlarza bronią. Jak ludzie wam mają ufać, w jaki sposób możemy skutecznie walczyć z pandemią, kiedy ludzie nie mają zaufania do władzy? Wtedy kiedy inni testowali w Europie na masową skalę, wy zajmowaliście się propagandą w telewizji publicznej. Wtedy kiedy trzeba było przygotowywać plany, wy zajmowaliście się walką z LGBT.

Ludzie wam nie ufają i dlatego dzisiaj jest tak, jak jest. Zapraszam panią posłankę Małgorzatę Tracz z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Debatujemy dzisiaj nad ustawami, o których powinniśmy byli rozmawiać już kilka miesięcy temu, kiedy już widzieliśmy, że jesienią czeka nas druga fala pandemii. Epidemii, która wbrew słowom rządzących nigdy tak naprawdę nie była w odwrocie i nie będzie do czasu upowszechnienia się szczepionki. Wasza ustawa jest przedstawiana przez wnioskodawców jako ustawa o dobrym samarytaninie, a tak naprawdę jest to ustawa o niczym innym jak o poborze do walki z epidemią. Ustawa ta daje wojewodom możliwość powołania do walki z epidemią studentów, doktorantów czy absolwentów, którzy jeszcze nie podeszli do egzaminów, oraz powołania osób, które nie podjęły pracy w zawodzie medycznym mimo posiadanego wykształcenia. I tu moje pytania do wnioskodawców: Czy będą jakieś konkretne zasady poboru osób z tej nowej grupy, z góry określona kolejność lub preferencje? Bo obecnie projekt tego nie precyzuje. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Michała Gramatykę z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Bardzo się cieszę, że uznali państwo jednak, że wirus jest groźny i że trzeba się go bać. Moje pytania dotyczą waszej filozofii działania, pewnej konsekwencji w tym działaniu. Zachowujecie się państwo trochę tak, jakby Ministerstwo Zdrowia było ministerstwem COVID-u. Jakie macie pomysły na innych pacjentów, na pacjentów onkologicznych, na pacjentów kardiologicznych? Co z tysiącami odwołanych planowych zabiegów i operacji? Dlaczego wasz nowy COVID-owy ład opiera się de facto na przenoszeniu, a wręcz kanibalizacji, zasobów pomiędzy jednym obszarem ochrony zdrowia a innym obszarem? Wczoraj pani posłanka Golbik i pan poseł Napieralski mówili o tym, jak zabieracie łóżka z psychiatrii dziecięcej i przenosicie je do COVID-u. W projekcie, który przedłożyli państwo, widać zapowiedź kolejnych kar. Kontrola, konsekwencja, kary - chełpił się jeden z waszych polityków. A może lepiej edukacja, motywacja, współpraca, zaufanie? Społeczeństwo jest waszym sojusznikiem w walce z tą pandemią. Warto w to uwierzyć. Dziękuję serdecznie. Zapraszam panią posłankę Iwonę Hartwich, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiaj chciałam upomnieć się o elektroradiologów. Proszę państwa, w ustawach, nad którymi pracujecie, przedstawiacie co chwilę nowe, zapominacie kompletnie o tej grupie medyków i pominięto właśnie tę grupę. Przypomnę: to osoby, które wykonują RTG, ale też różne inne badania. Te osoby są na pierwszej linii frontu w walce z COVID. Zwykle to do nich trafiają pacjenci z SOR i tam jest robiona diagnostyka. Minister zdrowia nigdy tych osób nie wymienia. Tam również są ludzie, którzy nie zdejmują COVID-owskiej odzieży. Im należy się tak samo wsparcie, jak innym grupom medycznym. Mam pytanie: Kiedy tej grupie zapewnicie należytą pomoc i ochronę? Dziękuję serdecznie. Zapraszam panią posłankę Monikę Rosę z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jak mówił pan minister Niedzielski, będzie jeszcze więcej, będzie jeszcze gorzej, będzie jeszcze trudniej. I najgorsze w tym wszystkim są działania pozorne - prężenie się na konferencjach prasowych, tworzenie pięknych obrazków na tle respiratorów czy przywiezionych na Stadion Narodowy łóżek. Te konferencje uspokajają wasze sumienia, ładnie wyglądają w telewizji publicznej, ale mają dla obywateli dramatyczne skutki. Powołują państwo w ustawie koordynatora ratownictwa medycznego. Ale co może koordynator, jeśli nie ma łóżek w szpitalach i brakuje lekarzy? Czy ten koordynator będzie decydował, kogo trzeba odpiąć od respiratora, kogo trzeba wyrzucić ze szpitala, a kto ma tam trafić? Czy będzie miał realny system, który pokaże mu, gdzie są wolne łóżka? Czy te wolne łóżka w ogóle będą? Szanowni państwo, poza koronawirusem istnieje jeszcze wiele innych chorób. Co z chorobami onkologicznymi? Co z chorobami serca? Co z innymi chorobami płuc, na które ludzie umierają codziennie? Miał być wielki plan powrotu do leczenia tych chorób, a przesuwane są zabiegi planowane. Ludzie się boją. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do odpowiedzi. Będziemy tych odpowiedzi mieli pięć, jeżeli wszyscy będą mieli ochotę zabrać głos. Zaczynamy od podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pana ministra Sławomira Gadomskiego. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan marszałek zapowiadał 30 pytań. Wydaje się, że pytań konkretnych padło tylko kilka, dosyć dużo krytyki i wolnych wniosków, ale niektóre bardzo cieszą. Rzeczywiście ja ze strony rządu deklaruję i odpowiadam na dużo tych postulatów dotyczących pracy merytorycznej.

Myślę, że ta otwartość z naszej strony deklarowana jest nie pierwszy raz, a mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mogli się przekonać, że jest ona faktem, bo dosyć wnikliwie przeanalizowaliśmy te projekty, które państwo złożyli, i nie są to rozwiązania, które negujemy. Co więcej, myślę, że rozwiązania te albo są już uwzględnione w ustawie złożonej przez posłów Prawa i Sprawiedliwości i zgodnej z tym, co wypracowywaliśmy wspólnie, albo są rozwiązaniami, które w inny sposób są już zaadresowane. Martwią mnie pewne sugestie co do tego, że z jednej strony mówimy: ministerstwo przespało, ministerstwo nie działa, ławy rządowe puste. Rząd jest zainteresowany tą dyskusją, pani poseł, i to, że w ławach rządowych siedzę tylko ja, a nie minister Niedzielski, nie zmienia faktu, że i jest zainteresowany, i wnikliwie przysłuchuje się tej dyskusji. Co więcej, myślę, że będziecie państwo mieli dzisiaj doskonałą okazję do tego, żeby zadać pytania zarówno panu ministrowi, jak i panu premierowi, bo taki porządek obrad został zaplanowany. Myślę, że w Komisji Zdrowia będziemy mieli znacznie więcej czasu, żeby można było do tych kwestii wrócić. Po raz drugi deklaruję: jesteśmy otwarci na rozsądne poprawki.

Nie różnicujemy ich dlatego, ponieważ minister zdrowia wydał Narodowemu Funduszowi Zdrowia polecenie, żeby we wszystkich szpitalach, które walczą z COVID, czyli wcześniej szpitalach jednoimiennych, a obecnie szpitalach trzeciego poziomu i drugiego poziomu, te dodatki były wypłacane. To nie jest polecenie nowe, nie jest to polecenie z dziś, to jest polecenie, które obowiązywało. A więc nie ma różnicowania, jest tylko wykazanie w ustawie wyjątkowego trybu w przypadku lekarzy czy personelu medycznego kierowanego przez wojewodów. Ale również ten personel, który walczy w tych szpitalach i jest tam zatrudniony na stałe, nie zmienia swojego miejsca, jest dodatkowo wynagradzany. Powiem więcej, Narodowy Fundusz Zdrowia czy fundusz COVID-owy, który jest w dyspozycji ministra zdrowia, wypłacił ogrom ekstraśrodków związanych właśnie z walką z COVID-em.

Poza tym już w przedstawionym Wysokiej Izbie projekcie ustawy budżetowej na następny rok w ogromnym stopniu zwiększyliśmy finansowanie inspekcji sanitarnej. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Panie ministrze, pozwoliłem panu jako marszałek Sejmu mówić minutę dłużej. Wie pan dlaczego? Dlatego że uznałem, iż sprawy istotne dla życia i zdrowia Polaków są najważniejsze. Wie pan, dlaczego mam taką refleksję? Bo gdyby tu siedział marszałek albo marszałkini z PiS-u, toby pan tej minuty nie dostał. A ja uważam, że sprawy najistotniejsze dla Polaków są ważne tak bardzo, że panu nie przerywałem. Dziękuję serdecznie.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Zacytuję wam biblijną Mądrość Syracha: w mowie jest albo sława, albo hańba. Druga sprawa. Oczywiście rozumiemy, że w takich sytuacjach zbójeckim prawem opozycji jest to, by krytykować, by nie mieć żadnej odpowiedzialności, mieć jakiś urobek populistyczny, demagogiczny, natomiast można się spierać, bo spór jest istotą demokracji, ale w innych kwestiach, na pewno nie o zdrowie i życie. Życie i zdrowie to jest sacrum, wszyscy powinniśmy je chronić i ratować. Natomiast wszelkie działania demagogiczne, populistyczne, kuglarstwo, sianie defetyzmu to nie w tym momencie, nie w tym momencie.

Jeden dzień zwłoki. To proszę się spytać ratowników medycznych, lekarzy na OIOM-ie, lekarzy na erce, co to znaczy.

Ponad 11 tys. zachorowań w 11-milionowych Czechach. Wszyscy spali? Przecież sytuacja jest dynamiczna, zmienia się z dnia na dzień. Trzeba reagować błyskawicznie. W medycynie dzień zwłoki to jest wieczność.

Rzeczywiście tam jest błąd techniczny, że uchyla się pkt 2b. Złożymy precyzyjną poprawkę.

Jeszcze raz przeczytam: na swój wniosek złożony do wojewody.

Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Zdzisława Wolskiego, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Straciliśmy ogromną ilość czasu.

Zamówiono ich nikczemnie mało.

Nie przeszkolono ich. Teraz już nie sposób ich przeszkolić, bo te, które mogłyby uczyć zawodu, są bardzo zajęte. Nie zrobiono nic. I to jest moja wielka pretensja pod adresem rządu.

Nawet nie ma na czym pracować, bo zatykają się laboratoria, punkty pobierania wymazów.

Zapraszam pana posła Szopińskiego, klub parlamentarny Lewica. Żałuję, że pan minister nie ustosunkował się do uwag, które przedstawiły Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wyraźnie napisała, i to jest uwaga do pań i panów posłów, którzy tutaj występują, że rejestry zgodnie z przepisami nie zawierają informacji o chorobach, ciąży lub posiadanym potomstwie. Nie są to informacje związane z wykonywaniem zawodu. Brak jest uzasadnienia odnośnie do gromadzenia takich danych. Należy podkreślić, iż informacje o stanie zdrowia są informacjami wrażliwymi i mogą być przetwarzane przez uprawnione organy na podstawie przepisów prawa. Tym samym naczelna rada pielęgniarek i położnych odpowiedziała na pytanie, jak ma się ten przepis do nakazania samorządom zawodowym medycznym w ciągu 7 dni przekazania wykazu osób, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Gdyby pan minister zechciał nakazać tym samorządom gromadzenie uwag i uaktualnienie takich danych, co oczywiście teoretycznie, legislacyjnie jest możliwe, to ów samorząd pielęgniarek i położnych powiedział, że zajęłoby mu to kilka miesięcy, a zatem byłaby to kwestia przyszłego roku. Zatem pytanie: Czy tędy droga? I ostatnia sprawa to jednodniowe opóźnienie. Otóż tak, musimy improwizować, bo zmarnowaliśmy czas. To, co się teraz dzieje, przypomina panikę. Ministerstwo Zdrowia nie zdało egzaminu. I teraz jest takie pytanie: Panie i panowie, kto to powiedział? Czy to padło z tej strony sali, czy z tej strony sali, czy skąd to padło? Otóż, rozwiązując tę zagadkę, powiem, że tak o tym wszystkim powiedział wasz poseł, panie i panowie z PiS, wasz poseł.

W związku z tym uwag o jednodniowe opóźnienie proszę nie kierować w tę stronę. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Dariusza Klimczaka, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Wysoka Izbo! Chciałbym podziękować w imieniu naszego klubu Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego - Kukiz15 za pozytywne ustosunkowanie się do przedstawionego przez nas projektu ustawy, który nazywamy premią dla bohatera. Właśnie dzisiaj podczas naszych obrad dostałem SMS od osób, których ta ustawa dotyczy, mianowicie dyplomowanych opiekunów medycznych. Właśnie ta grupa zawodowa często jest zapomniana, a wykonuje bardzo ciężką pracę od samego przyjęcia pacjenta do szpitala, po wszelkie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne, aż do samego końca, czasem jest niestety świadkiem ostatniego oddechu pacjenta. O tej grupie wiele osób zapomniało. Nie tylko premia dla lekarzy, nie tylko premia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, laborantów, ale także dla opiekunów medycznych.

Za to chciałbym podziękować, za te głosy z poszczególnych klubów, z wszystkich, bo nikt nie kwestionował słuszności tej propozycji. I mam nadzieję, że nasza propozycja będzie miała swoje odzwierciedlenie podczas prac komisji. Bo także chcielibyśmy, żeby był co najmniej ten zapis implementowany do dużej ustawy przedstawionej przez klub Prawa i Sprawiedliwości. Druga sprawa. Chciałbym, żebyśmy rzeczowo patrzyli na dyskusję, która toczy się w tej Izbie i która będzie się toczyła na posiedzeniach komisji i będzie miała swoją kontynuację w Senacie. Nie ma co się bulwersować, i mówię tutaj do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, z tego powodu, że opozycja w rzeczowy sposób krytykuje wasze działania bądź przypomina wasze zaniechania, które miały miejsce dotychczas. Uważacie, że za ostro ktoś na tej sali z opozycji potraktował wasze działania? To przypomnijcie sobie, kto powiedział, że opozycja jest gorsza od koronawirusa. Czy to nie był wasz przedstawiciel, prezydent Andrzej Duda, który wywodzi się z waszego środowiska? Tak.

Pierwsza nowelizacja po 5 latach? Tacy dobrzy jesteście dla sanepidu? Zmiany, które dotyczą nie systemu, a jedynie powoływania osób i odebrania kompetencji starostom - to zapewniliście sanepidowi, który dzisiaj oddycha rękawami?

To się już dzieje. Przecież każdy z nas dostaje do skrzynek mailowych uwagi od ratowników medycznych, w jaki sposób to powinno być rozwiązane - systemowo, a nie poprzez nakaz, nie poprzez decyzje. Co zrobi taki dyrektor szpitala czy ordynator, który ma oczywiście na sali dwa wolne łóżka, ale on przecież nie położy dwóch różnych jednostek chorobowych, gdzie jeden drugiego może doprowadzić do śmierci? I co, ten koordynator nakazem wrzuci taką osobę do szpitala? Przecież wy także macie, szczególnie w ministerstwie, sygnały z poszczególnych szpitali. Przecież naszymi uwagami, które tutaj zgłaszaliśmy, chcemy zmienić system funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Nie chcemy, żeby ilustracją służby zdrowia w Polsce były obrazki z Tarnobrzega, gdzie ludzie przychodzą pod parapet, biorą kije i uderzają, żeby ktoś im wydał receptę czy skierowanie. Chcemy, żeby tak wyglądał system ochrony zdrowia w Polsce? No chyba nie. Chcielibyśmy, żeby ten dostęp dla pacjenta był. A jeżeli nie potraficie tego zrobić w publicznym systemie ochrony zdrowia, dopuśćmy niepubliczny, prywatny system ochrony zdrowia, kilkaset szpitali, kilkaset gabinetów. Jeżeli nie mogę dostać się do publicznej ochrony zdrowia, niech państwo zapłaci za moje leczenie, kiedy pójdę do prywatnej.

Dziękuję serdecznie. Zapraszam do głosu pana posła Jacka Protasa z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan poseł Hoc rozpoczął od cytatu, więc pozwólcie państwo, że ja również zacytuję Fredrę, skieruję ten cytat do rządzących: „Niemała mądrość mądrze mówić, lecz największa - mądrze czynić” Słyszeliśmy z tej trybuny wiele pięknych słów, wiele zapewnień, natomiast jaka jest rzeczywistość, Polacy dzisiaj widzą. Zwrócę się również na początek do pana posła Piechy. Otóż, panie pośle, byłem dwie kadencje starostą, byłem dwie kadencje marszałkiem i zapewniam pana, że właścicielem szpitali powiatowych jest powiat, a właścicielem szpitali wojewódzkich - województwo. Szanowni Państwo! Padło pytanie o zaangażowanie samorządów terytorialnych w przeciwdziałanie pandemii.

Po drugie, samorządy województw zaangażowały ogromne środki, miliony w pomoc również dla przedsiębiorców, w granty dla tych, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, zarówno wykorzystując swoje środki, jak i w błyskawicznym tempie przesuwając środki europejskie na pomoc bezpośrednio przedsiębiorcom w walce z COVID-em. Kolejna sprawa, zakupy. Szanowni państwo, myśmy mieli spotkanie z nauczycielami i dyrektorami szkół przed 1 września. Otóż dyrektorzy szkół dostali z ministerstwa maseczki, które starczały dla szkoły na pierwszy tydzień funkcjonowania. I jak państwo myślą, kto w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach finansował zakup maseczek, środków dezynfekujących, wszelkiego innego sprzętu potrzebnego do tego, żeby chronić nasze dzieci, chronić nauczycieli, chronić rodziców? Samorządy terytorialne. Miliony złotych skierowano właśnie na ten cel. Szanowni Państwo! Trudno oszacować, jak wielkie koszty dopłat do transportu publicznego musi ponosić samorząd, jeżeli chce przewieźć swoich mieszkańców do pracy. Jednocześnie muszą być zachowane odległości. W autobusie, w pociągu może być określona liczba osób, natomiast te autobusy, te pociągi, to metro muszą się przemieszczać. Tego koszty ponosi samorząd terytorialny. Szanowni Państwo! Chcę powiedzieć, że rząd podejmuje kolejne decyzje, lepsze czy gorsze, trafne czy nie - najczęściej niestety, jak widzimy, z tą trafnością jest trudność - natomiast konsekwencje ponosi samorząd terytorialny.

To samorząd musi je przekładać na rzeczywistość, na codzienność, musi je sfinansować, zorganizować.

Dziękuję serdecznie. Zamykam dyskusję. Proponuję, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, aby Sejm skierował: - poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, zawarty w druku nr 683, - poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zawarty w druku nr 684, - poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zawarty w druku nr 685, - poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zawarty w druku nr 686, do Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Proszę państwa, ogłaszam przerwę do godz. 11.35. Dziękuję serdecznie.

Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19, a także wirusa grypy w czasie pandemii koronawirusa.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na początek chciałem przywołać słowa autorytetu medycznego, a zarazem osoby, która powinna nas wszystkich łączyć. Pan prof. Marian Zembala powiedział, że w obecnej sytuacji wszyscy powinni współpracować ponad podziałami. Nie ma innej opcji. To apel o solidarność. Apel o solidarność, język, który chyba wszyscy tutaj - niezależnie od różnic - rozumiemy. To właśnie ta solidarność w podejściu do epidemii mocno pomogła nam wiosną, bo równo 230 dni temu zaczęliśmy się zmagać z pandemią. Wysoka Izbo! Chciałbym tę moją informację skonstruować wokół sześciu głównych obszarów.

Po drugie, następnie powiem, co zrobiliśmy w ostatnich kilku miesiącach. Po czwarte, powiem o stanie gospodarki w czasie epidemii oraz o pewnych perspektywach gospodarczych. Po piąte, powiem o szkołach, o obostrzeniach, o poszczególnych branżach. Wreszcie po szóste, powiem także o naszej strategii i planach na przyszłość, w jaki sposób chcemy dalej walczyć z COVID-19.

Otóż niedawno, chyba dosłownie kilka dni temu, jeden z najbardziej uznanych periodyków medycznych na świecie, „The Lancet”, opublikował coś w rodzaju communis opinio doctorum, wspólnego zdania, konsensusu naukowego wszystkich tych, którzy zajmują się - i nie zgadzają często ze sobą, ale gdzieś jest też jakiś konsensus - COVID-19. Grupując to w pewne trzy obszary, można podkreślić, że chodzi tam o trzy podstawowe kwestie. Po pierwsze, jeśli chodzi o COVID-19, to najbardziej zabójcze są kontakt, bliskość, kontakt społeczny, częstość, mobilność społeczna, ponieważ one powodują przede wszystkim zakażanie się od siebie. Młodzi ludzie, którzy w mniejszym stopniu zakażają się w sposób groźny, jednocześnie są też bardzo dobrym, jak mówią epidemiolodzy, nośnikiem czy pasem transmisji koronawirusa do innych osób.

Otóż zgodnie z communis opinio doctorum jest to błędna teoria, ponieważ niezależnie od tego, że dość duża część populacji może ulec zakażeniu, co zresztą grozi również ogromną falą zgonów, to po drugie nie ma żadnej gwarancji, że za chwilę nie wybuchnie fala: ogniska, szerokie ogniska w różnych innych miejscach społeczeństwa, i że do tego taka strategia może prowadzić. Widzimy to po niektórych państwach. Przypomnijcie sobie strategię Szwecji czy Wielkiej Brytanii. To przecież na początku była darwinistyczna teoria odporności stadnej. Dziś widzimy po tej teorii, że ona nie działa tak, jak założyli sobie pierwotnie jej proponenci.

To jest coś, co przerywa transmisję w najbardziej skuteczny sposób. To dlatego dziś, jak porównujemy nasz stan łącznej liczby zachorowań do np. Włoch, to 50% więcej we Włoszech na milion mieszkańców, we Francji - 13 tys. [[Dzwonek]] na milion mieszkańców, w Polsce niecałe 5. Wreszcie w Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Holandii jeszcze dużo więcej.

I dzisiaj się również tej strategii trzymamy.

A więc z pewnymi fluktuacjami możemy mieć do czynienia jeszcze w dłuższej perspektywie czasu. Ale nasza strategia to przede wszystkim strategia i zasada: tak budować życie społeczne i gospodarcze, żeby móc uczyć się, pracować, żyć i jednocześnie nie zamykać gospodarki, jednocześnie przecinać ten pas transmisyjny COVID-19. Teraz przejdę do drugiego tematu, czyli co zrobiliśmy do tej pory, przez ostatnie miesiące. Przede wszystkim dokonywaliśmy ogromnych zakupów, i pokażę to na liczbach.

A więc w bardzo dużym zakresie te wszystkie materiały, które były potrzebne, dotarły do szkół w odpowiednim czasie.

Ile mamy dzisiaj możliwości testowych, szanowni państwo? Każdego dnia w ciągu lata zwiększaliśmy naszą wydolność i wydajność testów na koronawirusa.

W 2016 r. zatrzymaliśmy ten proces. Dzisiaj mamy możliwość testowania - zwększoną z 4 tys. do 80 tys. - 20 razy większą.

Strategia została wdrożona. W sierpniu, we wrześniu ona działała w taki sposób, jak spodziewaliśmy się, że zadziała. Natomiast we wrześniu pojawiło się bardzo wiele nowego ruchu, nowej mobilności społecznej. Zaraz o tym powiem, jak będę opisywał stan tu i teraz. Przygotowaliśmy również aplikację według najlepszych międzynarodowych standardów, aplikację STOP COVID.

Kupowaliśmy przede wszystkim sprzęt, który leczy najciężej chorych na koronawirusa, czyli respiratory. Respiratorów kupiliśmy tyle, że potroiliśmy stan łóżek z respiratorami między sierpniem a dniem dzisiejszym.

Tak więc wszystkie szpitale, każdy, niezależnie od tego, jaki jest organ założycielski, czy marszałkowski, czy miejski, każdy, który chce podłączyć respirator, dostanie ten respirator, ponieważ mamy dzisiaj wolnych respiratorów blisko 3 tys. To jest skutek myślenia strategicznego w miesiącach letnich, kiedy wiedzieliśmy, że możemy się zderzyć z większą liczbą zapotrzebowania na respiratory.

Jednocześnie też w całej strukturze szpitalnej zmienialiśmy przyporządkowanie w taki sposób, żeby odpowiedzieć na wyzwania, z którymi się mierzymy. Powiem o stanie w dniu dzisiejszym, gdzie jesteśmy tu i teraz, czyli jest to trzecia część mojego wystąpienia, mojej informacji.

To duży procent, ale cały czas zwiększamy bazę łóżkową. Wyszliśmy ze stanu, jak powiedziałem, 6 tys. łóżek jeszcze 6 tygodni temu, 7 tygodni temu, dzisiaj jest to 16, 17 tys. łóżek.

Ale duża liczba zakażeń, 9, 10 tys. zakażeń, którą musimy zatrzymać, jednocześnie oznacza, że musi rosnąć liczba łóżek dostępnych dla pacjentów. W naszym planie, o którym powiem w ostatniej części mojej wypowiedzi, jest założenie co najmniej kolejnych 15 tys. łóżek. 13 tys. już jest zidentyfikowanych w szpitalach powiatowych, w szpitalach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej, MSW czy Ministerstwu Zdrowia.

To spowodowało z pewnym opóźnieniem - bo epidemia działa z odłożonym skutkiem: 2–3-tygodniowym, czasami trochę szybciej - że zaczęła pojawiać się większa liczba osób zakażonych i już nie w takim układzie ognisk, układzie ogniskowym, jak to było wiosną, tylko jest to szeroko rozpowszechnione w całym społeczeństwie. Żeby to przerwać, co teraz, tu i teraz zrobiliśmy? Na początku października wdrożyliśmy nowe obostrzenia, obowiązek noszenia maseczek przez wszystkich. Jeszcze do tego wrócę w piątej części mojej wypowiedzi, bo wiem, że są sceptycy także tutaj, na sali. Ale kierujemy się badaniami, opiniami ekspertów, wirusologów i dlatego to zaleciliśmy. Dzięki temu nastąpiła zmiana, którą w badaniach naukowych określa się mniej więcej jako poziom: 13% mniejszy wskaźnik R, czyli ten wskaźnik, który w sposób poziomy pokazuje, jaka jest transmisja z człowieka na człowieka w całej populacji. Co zrobiliśmy następnie? Następnie posłużyliśmy się kolejnymi badaniami naukowymi dotyczącymi szkół.

Czyli znowu poprzez ten nasz ruch we właściwym kierunku, który ogłosiliśmy w zeszłym tygodniu, mamy krok w kierunku ograniczenia transmisji społecznej. To być może dlatego jeszcze tydzień temu niektórzy się obawiali, że będzie kilkanaście tysięcy zakażeń. Tyle nie ma, ale my zakładamy najgorszy scenariusz. Dlatego będziemy na pewno tworzyć taki system szpitalnej dostępności łóżek dla chorych na COVID-19, żeby nie spotkało nas to, co spotkało Europę Zachodnią, spotkało najbogatsze kraje świata - tak można śmiało powiedzieć - czyli: nie leczymy pacjentów powyżej pewnego poziomu wieku. Pamiętacie to państwo: w Hiszpanii, we Francji, w Belgii.

Nie mamy sytuacji takiej jak w niektórych krajach Europy Zachodniej, gdzie ta liczba jest daleko bardziej wykorzystana. Jeśli chodzi o nasze możliwości testowe, dziś to była jedna z wyższych liczb testowych, 51 czy 51,5 tys. Ale były już dni, kiedy testowaliśmy ponad 60 tys. pacjentów, ponad 60 tys. Polaków. Nasze możliwości, moce wydajnościowe całego systemu testowania są więc wyższe już dzisiaj i cały czas podnoszone tak, żeby w sytuacji kiedy trzeba będzie testować więcej, można było testować więcej. A więc nasza strategia, nasza droga środka - kiedy odrzucamy jedno ekstremum, czyli tych, którzy są przeciwnikami jakichkolwiek obostrzeń, ale także tych, którzy chcą zamknięcia gospodarki, natychmiastowego zamknięcia wszystkiego, tak jak wiosną albo jeszcze bardziej - jest najbardziej właściwa, dlatego że my musimy w dłuższym horyzoncie czasowym nauczyć się żyć z pandemią, ponieważ ona może słabnąć i może się ponownie wzmagać. Dlatego musimy z całą mocą zaadaptować takie metody, które doprowadzą do tego, że będziemy uczyć się pewnie zdalnie w większości - jeszcze do tego wrócę - będziemy pracować, będziemy po prostu żyć, ale będziemy chronić naszych seniorów, naszych najsłabszych, będziemy mogli leczyć wszystkich ludzi, którzy będą tego leczenia potrzebowali. To jest nasza strategia na tu i teraz i z tego punktu wyjścia w ostatniej części opowiem o naszych planach na przyszłość. Teraz kilka słów w czwartym punkcie, o gospodarce. Otóż, szanowni państwo, to, co spotkało gospodarkę świata, gospodarkę Europy, nie było zapisane w żadnych podręcznikach ekonomicznych. Nikt nigdy nie mierzył się z takimi problemami. Najpierw kompletny szok, tzw. asymetryczny szok podażowy, asymetryczny szok popytowy, pełne zahamowanie mechanizmów płynnościowych w gospodarce. Na to wszystko zareagowaliśmy błyskawicznie, zareagowaliśmy tarczą finansową, zareagowaliśmy tarczą antykryzysową, poduszką płynnościową dla przedsiębiorców, która cały czas tam jest. Mierzona obiektywnymi wskaźnikami - ta poduszka jest i według finansistów, ekonomistów wystarczy jeszcze na kilka miesięcy. Wiem, że są branże, które są i będą dotknięte bardziej. O tym jeszcze parę słów za chwilę powiem. Nie było żadnych rad w żadnych podręcznikach, ani Keynesa, ani Krugmana, ani Friedmana, ani Hayeka, ani innych wielkich ekonomistów, jak poradzić sobie z takim kryzysem. Przeszliśmy przez to relatywnie suchą stopą. ponieważ we wskaźnikach OECD, we wskaźnikach Komisji Europejskiej, w tych 2 latach Polska ma szansę przejść najbardziej suchą stopą przez te bardzo wzburzone wody, również tej drugiej fali. Tej drugiej fali, o której pan przewodniczący Koalicji Obywatelskiej mówił, że jesienią to już pandemia będzie w zaniku, bo takie macie ekspertyzy. Na marginesie: niech pan pokaże te ekspertyzy, panie przewodniczący. A więc, szanowni państwo, dalej. Gospodarka. Co najlepiej świadczy o tym, w jaki sposób gospodarka przechodzi przez ten największy kryzys od ok. 100 lat? Otóż miarą tego, w jaki sposób przechodzimy kryzys, jest to, czy udaje się utrzymać miejsca pracy. Poprzez nasze tarcze finansowe utrzymaliśmy 5 mln miejsc pracy. To wielkie osiągnięcie, które doprowadziło do tego, że Polacy dzisiaj mogą mimo tych ogromnych zagrożeń gospodarczych spać spokojniej niż wielu innych obywateli Europy. Ostatnio międzynarodowy fundusz podał dane, że nasza odpowiedź fiskalna, budżetowa była największa w Europie. Mówiliście z jednej strony: wydatki za małe, a z drugiej strony: deficyt budżetowy za duży. No to jest żelazna logika, rzeczywiście.

Ten deficyt jest, ale dzięki temu ochroniliśmy miejsca pracy. Bo trzeba zdać sobie z tego sprawę, że zależność między epidemią a gospodarką jest bardzo duża, korelacja jest ogromna i jednocześnie ta wzajemność jest dwustronna. Im szybciej uda nam się zwalczyć epidemię, im ona mniej atakuje, tym gospodarka czuje się w takiej sytuacji lepiej, tym perspektywy przed gospodarką są lepsze. Ale także w drugą stronę: jeżeli jest tąpnięcie gospodarcze, jeżeli jest w gospodarce rosnące bezrobocie, gwałtownie rosnący dług publiczny, gwałtowny spadek PKB.

W Wielkiej Brytanii - minus 22% w II kwartale. My przechodzimy przez to inaczej i to jest najlepsza miara, relatywna, miara porównawcza, w jaki sposób ratujemy miejsca pracy, w jaki sposób ratujemy przedsiębiorców przed bankructwem, ratujemy ich udział w rynku. I wy wiecie, że ta tarcza jest dobra. Wy wiecie, że ona działa, bo tutaj w Sejmie pan przewodniczący Budka i pan prezes Kosiniak-Kamysz w rozmowie mówili o tym.

A więc powiem ostrożniej: będziemy w pierwszej trójce albo w pierwszej piątce całej Unii Europejskiej. I to jest miara skuteczności działań gospodarczych Prawa i Sprawiedliwości. Teraz przejdę do tego piątego obszaru, który chciałem omówić: szkoły, obostrzenia, branże. A więc, po pierwsze, kwestia szkół. Tutaj trzeba zacząć od tego, że w epidemii. Nie ma takich miejsc w sytuacji szeroko rozprzestrzenionej epidemii, które są całkowicie bezpieczne dla kogokolwiek. Bo epidemia rzeczywiście ma już dzisiaj charakter poziomy, horyzontalny, rozprzestrzeniła się wszędzie w społeczeństwie. Dlatego kierujemy się zdaniem ekspertów i na początku zamknęliśmy dla nauki stacjonarnej szkoły średnie, szkoły ponadpodstawowe, ponieważ to jest ponad 1,5 mln osób, uczniów, którzy tworzą ten ruch społeczny, tworzą mobilność i powodują, że liczba kontaktów społecznych jest większa.

A to dlatego, że zdaniem ekspertów i epidemiologów - chociażby proszę przeczytać czy posłuchać tego, co mówi profesor Gut - dla osób do 9. roku życia zakażenie raczej bardzo, bardzo rzadko skutkować może bardzo poważnymi konsekwencjami dla zdrowia. Natomiast już u nastolatków to ryzyko rośnie, aczkolwiek też na szczęście u nastolatków powikłania są bardzo rzadkie. To dopiero osoby starsze musimy chronić za wszelką cenę i doprowadzić do tego, żeby tam, w tej grupie było najmniej kontaktów społecznych. Dlatego, drodzy państwo, przeznaczyliśmy w pierwszej części, i także latem, tworząc przestrzeń techniczną do nauki zdalnej, 370 mln zł, a teraz przeznaczamy kolejne 300 mln zł na naukę zdalną dla szkół. Bo z drugiej strony trzeba powiedzieć wprost i szczerze, że nauka zdalna to jest dalece nie to samo, co nauka stacjonarna. Nauczyciel zawsze jest w stanie lepiej przekazać wiedzę w trybie stacjonarnym, dlatego rozumiem nauczycieli i rozumiem też tych wszystkich, którzy woleliby taki tryb nauczania. Ja też bym wolał. Ale musimy jednocześnie odpowiadać na to, co grozi nam, a grozi nam przyrost liczby osób zakażonych i ten przyrost chcemy hamować, tak żeby za jakiś czas on również spadał. A więc szkoły będziemy w takim cyklu reorganizować. I miejmy też na uwadze to, że dla dzieci najmłodszych, dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym do 9., 10. roku życia, zdaniem psychologów, psychiatrów dziecięcych nauka w klasie, w szkołach jest również bardzo ważna ze względu na efekty społeczne, nie tylko efekty edukacyjne, pedagogiczne. Dlatego staramy się to różnicować. Teraz, szanowni państwo, są tacy fałszywi apostołowie antymaseczkowi, którzy wzywają wszystkich do tego, żeby nie nosić maseczek. O siebie się boją, a o innych nie troszczą się w takim samym stopniu. Mamy więc do czynienia z pewnego rodzaju obłudą. Poprzez te wszystkie obostrzenia, wszystkie rady, które dają nam grupy ekspertów, chcemy doprowadzić do tego, żeby ta transmisja, ten współczynnik R był odpowiednio mniejszy, odpowiednio niski. Dlatego właśnie podkreślamy, że te obostrzenia muszą być rygorystycznie przestrzegane.

To jeszcze można włączyć do tej części, w której mówiłem o tym, co działo się w ostatnich miesiącach. Otóż nasze służby mundurowe skontrolowały 20 mln osób, które znajdowały się na kwarantannie. 20 mln telefonów, wizyt, stukania do drzwi.

Jest to potrzebne, żeby każdy z nas trzymał się tych przepisów. Żyjemy nie tylko dla siebie.

Ale chcemy, jak powiedziałem wcześniej, uczyć się żyć, pracować i korzystać z usług różnych branż w taki sposób, który byłby bezpieczniejszy.

Dlatego chcemy to doregulować, jeśli mogę tak powiedzieć, czy wzmocnić tę regulację również na poziomie ustawowym. I za współpracę w tym zakresie również dziękuję. Szanowni Państwo! To wypośrodkowanie jest potrzebne, żeby z jednej strony ochronić jak najwięcej ludzi, a z drugiej chronić miejsca pracy, by nie doszło do tąpnięcia gospodarczego. Dlatego przejdę teraz do naszej strategii na przyszłe miesiące, może nawet na przyszłe kwartały. Na czym ona polega? Otóż mamy trzy główne cele tej strategii. Po pierwsze, ochrona zdrowia, ochrona systemu zdrowia i ochrona służby zdrowia, czyli ochrona tego, co stoi u podstaw służby społecznej w celu zmniejszania zagrożenia COVID-19. Po drugie, ochrona gospodarki, ochrona miejsc pracy. I po trzecie, ochrona seniorów, najsłabszych, ponieważ największa liczba zgonów jest właśnie w tej grupie, a więc wiele naszych działań - za chwilę powiem o niektórych - odnosi się do tego obszaru.

Ona już uratowała ileś istnień ludzkich. Jednocześnie te działania będą ewoluowały, ponieważ epidemia jest groźna również przez to, że jest nieznana, jest zjawiskiem nieokiełznanym, nieprzewidywalnym. A co to oznacza? Dla każdego stratega to oznacza, że nasza reakcja musi być elastyczna. Musimy zakładać sobie bufor elastyczności, pewien bufor, i on tutaj jest wkomponowany. I teraz o nim powiem w kontekście drugiej, trzeciej i czwartej linii obrony. Druga linia obrony to nasz system ochrony zdrowia, to nasze już dzisiaj 16 tys. łóżek szpitalnych, 40% więcej niż jest dzisiaj wykorzystywanych.

Trzecia linia obrony to tworzenie dodatkowych 13 tys. łóżek szpitalnych wraz z odpowiednią proporcją podłączeń respiratorowych, podłączeń tlenowych. Przypomnę, że tylko w ostatnim tygodniu rozdystrybuowaliśmy 350 respiratorów do szpitali i 300 kardiomonitorów. A więc tworzenie dodatkowych łóżek szpitalnych z zasobów MON, MSW, Ministerstwa Zdrowia, szpitali powiatowych, w których dokonujemy pewnej reorganizacji. To nas doprowadzi do poziomu ok. 30 tys. łóżek, łóżek przeznaczonych tylko dla pacjentów z COVID-19. To nas doprowadzi do ok. 30 tys. Drodzy rodacy, żeby jednak czuć się jeszcze bardziej bezpiecznie, tworzymy czwartą linię obrony. To są te szpitale tymczasowe, tak je nazywamy. To są szpitale w hali Expo, na stadionie, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W każdym województwie chcemy mieć tego typu zasoby łóżkowe dodatkowo.

To jest nasza czwarta linia obrony i oby ona nie została wykorzystana. Teraz to, co dodatkowo świadczy o naszym myśleniu strategicznym, o myśleniu do przodu.

A więc myślimy już o tych, którzy doznają, którzy mogą doznać uszczerbku na zdrowiu, i będziemy ich rehabilitować, leczyć. To jest ośrodek w Głuchołazach. A więc już jest pilotaż, który działa, który jest czynny, który przecież musiał być przygotowany w miesiącach letnich. Dzisiaj tę strategię będziemy proliferować, będziemy rozprzestrzeniać na inne ośrodki, bo niestety COVID-19 to choroba groźna.

To nie jest właściwa strategia. Następny obszar, wątek, o którym wspomniałem, że go rozwinę w dwóch zdaniach - Korpus Wsparcia Seniorów. Jutro lub pojutrze, w najbliższych dniach przedstawię, w jaki sposób Korpus Wsparcia Seniorów będzie działał. Proszę was o to, nasi dziadkowie i babcie, nasi rodzice, nasze mamy, ojcowie. Ci, którzy nie pracują, którzy mogą pozostać w domu - jeśli możecie pozostać w domu, zostańcie. Skontaktujcie się z odpowiednimi służbami, one pomogą w dostarczeniu żywności, lekarstw czy innych artykułów pierwszej potrzeby. Korpus Wsparcia Seniorów doprowadzi do tego. I to jest bardzo ważna część naszej odpowiedzi, naszej strategii na przyszłość. Kolejna kwestia, którą rozwijamy, to ciągłe czerpanie z doświadczeń innych. krajów europejskich, które podpisały umowę, razem z Komisją Europejską, z siedmioma bądź ośmioma, dzisiaj już chyba ośmioma, firmami farmaceutycznymi, największymi firmami świata, które pracują nad szczepionką, po to, żeby być w pierwszej grupie, jeżeli szczepionka zostanie wynaleziona, tych, którzy mogą z tej szczepionki skorzystać.

Dziękuję za przypomnienie. Panie pośle, szczepionki na grypę - mamy dzisiaj, już zakupionych i zamówionych, ponad 3 mln szczepionek.

Mało tego, dla seniorów powyżej 75. roku życia, a chcę, żeby to było powyżej 70. roku życia, szczepionki te będą dostępne bezpłatnie po to, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo skumulowania się tych chorób. To jest nasza strategia, to jest myślenie na przyszłość. Strategia, która zakłada te cztery linie obrony przed COVID-19. I teraz, szanowni państwo, na zakończenie. Idziemy tą właśnie drogą środka. Z jednej strony mamy tych, którzy chcą doprowadzić do całkowitego lockdownu, którzy wzywają do jak największych. Z drugiej strony mamy tych, którzy chcą zignorować COVID-19. Ale przestrzegam. Może doprowadzić do tego, że zamknięcie, lockdown gospodarki, części gospodarki, będzie dłuższy, głębszy i z większymi skutkami gospodarczymi. Dlatego ta droga środka jest tak potrzebna. Odrzućmy ten dziwny sojusz skrajnych negacjonistów i tych, którzy proponują natychmiastowe zamknięcie gospodarki, podobnie jak część naszych oponentów również w Sejmie.

Dlatego warto, żeby ponad podziałami, w duchu solidarności walczyć z COVID-19. Musimy nastawić się na dłuższą walkę. Może będzie kolejna fala, może będzie szczepionka. Tego dzisiaj nie wiemy. Kto nie popełnia błędów, niech pierwszy rzuci kamieniem. Zrobimy wszystko, żeby bronić naszych seniorów, chronić gospodarkę i służbę zdrowia, chronić zdrowie i życie wszystkich naszych obywateli. Szanowni Państwo!

Epidemia w końcu - jak ogromna większość epidemii czy wszystkie epidemie - zostanie przez człowieka w skuteczny sposób zwalczona, ale musimy jednocześnie ochronić miejsca pracy, możliwość świadczenia pracy i naszą gospodarkę.

Tą szczepionką jest solidarność. Dziękuję bardzo.

Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Dzisiejsze wyniki mówią same za siebie - 10 tys. nowych zakażeń.

Chcę państwa zapewnić, że mamy świadomość różnych wariantów, różnych scenariuszy, również tych najczarniejszych, które zakładają wykładniczy przyrost liczby zachorowań, dlatego przygotowujemy się na każdy scenariusz.

To jest nasza gwarancja bezpieczeństwa.

Bardzo się cieszę, że mogę z tego miejsca powiedzieć, że również sektor prywatny włączył się w walkę z COVID-em. Jestem po rozmowach z przedstawicielami prywatnych szpitali, prywatnych jednostek lecznictwa. Mamy deklarację, wraz ze wskazaniem konkretnych lokalizacji, co do blisko 1 tys. dodatkowych łóżek. Ten 1 tys. może nie robi wrażenia, ale proszę pamiętać, że prywatna służba zdrowia w Polsce, mówię o tym poziomie szpitalnictwa, to blisko 4 tys. łóżek, czyli prywatna służba zdrowia zadeklarowała blisko 25% swoich zasobów na walkę z COVID-em. To jest wielkość porównywalna z tą, o której mówił pan premier, którą chcemy osiągnąć również w sektorze publicznym. Tutaj będziemy chcieli mieć w tym pierwszym ruchu mniej więcej 30 tys. łóżek, a potem ze szpitali tymczasowych - kolejne tysiące. Szanowni Państwo! Jeżeli patrzymy na przebieg pandemii tak naprawdę od początku, od marca. Pan premier mówił o strategii, ja zejdę piętro niżej i powiem kilka słów o taktyce. Mamy naprawdę co najmniej trzy wyraźne okresy przebiegu tej pandemii.

Potem weszliśmy we wrzesień. Wrzesień już niestety okazał oblicze drugiej fali i mieliśmy do czynienia ze wzrostem, ale nie aż tak dynamicznym, bo miał on charakter liniowy. Przypomnę państwu, że na początku września liczba zachorowań wynosiła dokładnie 550, a na koniec września mieliśmy liczbę zachorowań wynoszącą 1500, czyli wrzesień spowodował już potrojenie się liczby przypadków. Wtedy, w pierwszych dniach października, niestety ten trend się zmienił - na trend wykładniczy. Ten przyrost już nie był taki stopniowy, systematyczny, tylko mieliśmy do czynienia z dużym przyspieszeniem tempa rozwoju pandemii. Przypominam, że w październik wchodziliśmy z liczbą zakażeń 1500, podczas gdy dzisiaj mamy wynik 10 000. To oznacza sześciokrotny przyrost, a miesiąc się jeszcze nie skończył. Dlatego w zależności też od typu, od przebiegu tej pandemii dobieraliśmy odpowiednie środki. Mówimy o wakacjach. Rozbudowaliśmy rezerwy. To jest nieprawda, chociażby ze względu na to, że w wakacje staraliśmy się przywrócić dostępność służby zdrowia, która została na samym początku praktycznie zamrożona.

A więc tym bardzo ważnym zadaniem, które było realizowane w tych letnich miesiącach, było przywrócenie dostępności w tych zakresach, które zostały zamrożone w pierwszych dniach pandemii.

Wprowadziliśmy rozwiązanie, które polegało na tym, że lekarze rodzinni będą mogli zlecać badania. Na początku chcieliśmy mieć taki wymóg po badaniu fizykalnym, ale potem w dialogu z lekarzami rodzinnymi wypracowaliśmy rozwiązanie, które jest oparte na ankiecie, odwołuje się do nowoczesnej wiedzy. Proszę zobaczyć, jakie są efekty. On jest też efektem powiększania tzw. zdolności laboratoriów do wykonywania badań. To było robione w wakacje, to było robione właśnie w czasie letnim. Mieliśmy już kilka dni, kiedy te 60 tys. było przekroczone. Z jednej strony to się bierze z rozbudowy, ale z drugiej strony to jest bardzo poważna zasługa lekarzy rodzinnych, którym bardzo dziękuję z tego miejsca za włączenie się w proces leczenia - już nie tylko zlecania testów, bo we wrześniu również wypracowaliśmy rozwiązanie, w ramach którego pacjenci skąpoobjawowi bądź bezobjawowi są kierowani na izolację bądź prowadzeni podczas tej izolacji przez lekarzy rodzinnych. Czyli mamy i większą testowalność, lepsze rozeznanie, gdzie jest ten wirus.

Szanowni Państwo! To włączenie POZ-etu i strategia testowania, myślę, pozwalają nam wiedzieć, z jakim naprawdę problemem mamy do czynienia. Sytuacja jest bardzo poważna i dlatego też podejmujemy drastyczne środki. Drastyczne środki, które dotyczą obostrzeń i które są z naszego punktu widzenia hamulcem rozwoju wykładniczego pandemii. Ten hamulec musimy nacisnąć wszyscy bardzo mocno, bardzo dynamicznie, bo tutaj mamy obostrzenia, pan premier zapowiedział, że dzisiaj będą dalsze zaostrzenia, ale w tej chwili rzeczywistość wygląda tak, że my na bieżąco monitorujemy liczbę tzw. czerwonych stref, ta liczba dochodzi już do 300 przy liczbie powiatów wynoszącej 380. A więc musimy ten hamulec nacisnąć, musimy zwiększyć obostrzenia, bo bronimy nie tylko bezpośrednio zdrowia ludzi, ale bronimy też wydolności systemu opieki zdrowotnej, bo nie ukrywajmy, że w tej chwili testujemy tę wydolność. Szanowni państwo, przejście z liniowego charakteru wzrostu liczby dziennych zachorowań na charakter wzrostu wykładniczego wymaga od nas działań, wymaga działań związanych z wprowadzaniem obostrzeń, stosowaniem pewnej zasady odpowiedzialności społecznej - wyrazem tego, czy jestem egoistą, czy jestem altruistą, jest z mojego punktu widzenia w tej sytuacji noszenie maseczki, stosowanie innych reguł życia społecznego, bo one już powinny mieć status reguł życia społecznego, czyli dystans, czyli dezynfekcja, czyli stosowanie również aplikacji, która jest do tych celów dedykowana, dostępna za darmo we wszystkich sklepach internetowych, mobilnych, ona jest zresztą oparta na rozwiązaniu, które funkcjonuje w Niemczech.

Dlatego przygotowaliśmy pakiet rozwiązań legislacyjnych i mam nadzieję dzisiaj - przy otwartości na dyskusję w komisji, którą deklaruję - chciałbym, żeby dzisiaj stał się on kolejnym orężem walki z pandemią, orężem, który pozwoli nam dać większe gwarancje bezpieczeństwa personelowi, większą motywację finansową i poprawić warunki pracy, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo pacjenta. Ja na razie nie będę tutaj mówił o wszystkich szczegółach, bo tak jak powiedziałem, ostateczny kształt ustawy na pewno będzie wypracowany po pracy w komisji, bo pierwsze czytanie mamy już za sobą. Ale bardzo proszę, i zwracam się tu z pozycji wszystkich pacjentów i medyków, bardzo proszę o współpracę, bardzo proszę o życzliwe spojrzenie na rozwiązania, które proponujemy. Bardzo proszę o współpracę. Dziękuję, panie ministrze.

Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Bolesław Piecha, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam przedstawić stanowisko dotyczące informacji pana premiera o stanie przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i w konsekwencji choroby COVID-19, a także tej sytuacji, gdy mamy jednak sezonowość zachorowania na grypę. Muszę powiedzieć, że z 5-letnią przerwą prawie 20 lat zasiadam w tej Izbie i rzadko się słyszy tak merytoryczne, tak szczere i z taką dużą pokorą wystąpienie pana premiera, oparte głównie na faktach - nie na domniemaniach, nie na jakichś różnych przykładach sprzecznych czy skrajnych, ale na tym, co dokładnie dzisiaj wiemy.

To jest bardzo ważne. Istnieje w przestrzeni publicznej wiele różnych dziwnych zjawisk i dziwnych komentarzy. Jak kiedyś każdy Polak znał się na ochronie zdrowia, tak dzisiaj wszyscy znają się na epidemiologii, wszyscy wiedzą, co to jest wirus COVID, co to jest choroba COVID-19, wszyscy mają. odpowiednie recepty. Ja zawsze wysłuchuję oczywiście w tej sali tzw. sejmowych krzykaczy, którzy różne podpowiadają wieści, ale sądzę, że to przemówienie, to wystąpienie było bardzo dobre. Co zrobiliśmy - wiemy. Zrobiliśmy to, na co był przygotowany świat. Świat nie znał i nie zna rozwoju tej epidemii, ponieważ żadne państwo na świecie. żadna instytucja naukowa, żaden instytut dzisiaj nie wynalazły środków, które zapobiegają epidemii, czyli szczepionki, bo to na szczepieniach ochronnych opierało się w historii medycyny zapobieganie epidemiom, ani nie wynalazły lekarstwa i - trudno, będę sceptykiem - szybko go nie wynajdą, ponieważ 60 albo 70 lat znamy budowę wirusa i nikt leku na wirusa do dzisiaj nie wymyślił. A była i Ebola, a był i AIDS. Nadal nie mamy leku na tego typu wirusy i pewnie na tym się musimy dzisiaj opierać. Pan premier powiedział, jakie były strategie, a pan minister uzupełnił o to, co się stało na przełomie września i października. Znowu też nikt prawdopodobnie z ekspertów w tym konsensusie naukowym nie zakładał, że akurat te pierwsze miesiące, te dni wrześniowo-październikowe będą szczytem epidemii. To jest sezon grypowy. W związku z tym elastycznie trzeba podejmować różnego rodzaju działania i o tych działaniach pan premier z dużą odwagą i z dużą pokorą powiedział, bo tylko ten może krzyczeć, kto nie zna słowa: pokora i uważa, że siły natury, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, są pod pełną naszą kontrolą. Być może są tacy na sali, ale oni opierają się o tzw. idee nadwartościowe, a to już jest przyczynek do badań psychiatrycznych. Chciałbym powiedzieć, że ważną sprawą są obostrzenia, które my wszyscy odczuwamy.

Nie wiem dlaczego. Ale chodzę w tej maseczce, ponieważ jest to pierwszy etap możliwości postawienia bariery dla szerzenia się tego wirusa.

A więc te obostrzenia w tym wymiarze społecznym muszą istnieć. Drugim rodzajem obostrzeń oczywiście są takie obostrzenia, które wzmacniają ten nasz dystans społeczny i one dotyczą kwestii również takich, żeby gospodarka oczywiście nie ucierpiała albo jak najmniej ucierpiała, żeby po prostu nie ucierpiała, bo my się musimy rozwijać. My jesteśmy społeczeństwem, które ma swoje aspiracje, ma swoje oczekiwania i te oczekiwania musimy realizować, a istotą, czyli sensem i możliwością realizacji tych naszych oczekiwań, zamierzeń jest praca i miejsca pracy są istotnym elementem obrony przeciwko fatalnym skutkom pandemii. Chciałbym również powiedzieć o tym, co jest robione, i to być może w przyspieszonym czasie. To jest przygotowanie infrastruktury szpitalnej do tego, żebyśmy mogli chorym, zakażonym po prostu profesjonalnie i z pewną godnością się zaopiekować. Pan premier powiedział wyraźnie, że najpierw chodzi o przystosowanie pewnych oddziałów, pewnych łóżek szpitalnych w szpitalach wojewódzkich, w szpitalach klinicznych, w szpitalach powiatowych, a dopiero w ostatniej kolejności o przygotowanie tzw. szpitali tymczasowych, przez niektórych nazywanych szpitalami polowymi. Również jesteśmy przygotowani - i to bardzo ważna rzecz - jeżeli chodzi o sprzęt dla najciężej chorujących, czyli respiratory. Nie każdy potrzebujący tlenu musi być od razu przyłączony do respiratora. To są namioty, to są instalacje tlenowe.

Jest to też bardzo ważne, żeby podmioty tworzące szpitale: wojewodowie, marszałkowie, starostowie, współpracowali z rządem przy tworzeniu tej strategii. Ostatnią sprawą, o której chciałbym powiedzieć - i to jest również bardzo ważna rzecz - mówiłem o tym 3 godziny temu w czasie omawiania tej ustawy, która powoduje również mobilizację tego, co jest istotą przeciwdziałania i leczenia chorób, jest kadra pracowników medycznych. Zostali oni docenieni i to w sposób bardzo wyraźny. Ja chyba w tej 20-letniej historii nie słyszałem o podwyżkach 200-procentowych, o tym, żeby tak mocno dohonorować ludzi, którzy walczą z epidemią. Nie słyszałem również o tym, żeby łamać albo zmieniać przepisy ZUS-owskie tak, że oni mają całkiem inne świadczenia, jeżeli ulegną zakażeniu lub będą musieli być na kwarantannie, a to nie znaczy, że ulegli zakażaniu. Tam też trzeba wprowadzić środki finansowe i te środki są oczywiście ZUS-owskie. Również trzeba powiedzieć, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy, że te zadania będą wprowadzane w dialogu. I to nie jest prawdą, że ktoś kogoś będzie gdzieś zmuszał, ale sądzę, że po drugiej stronie społecznej, po drugiej stronie, czyli chodzi o pracowników ochrony zdrowia, jest pełna zgoda. My, lekarze, jesteśmy powołani - nie przymuszani - do leczenia chorych i pewnie z tego się wywiążemy. Panie Premierze!

Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Borys Budka, Koalicja Obywatelska.

Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Panie Premierze! Wreszcie odważył się pan stanąć przed nami po wielu miesiącach apeli, próśb, by problem pandemii traktować poważnie i ponad podziałami politycznymi. Unikaliście tej debaty, bo zajmowaliście się samymi sobą. Walczyliście o stołki, wpływy, dzieliliście pieniądze. Nawet w ostatnich dniach urzędowania potrafiliście wypłacać pracownikom rekordowe nagrody, a Polaków zostawiliście samych. Dziś padł kolejny rekord zachorowań - ponad 10 tys. przypadków, 130 osób zmarło. Ludzie nie potrafią dodzwonić się do sanepidu. Szkoły nie wiedzą, co mają robić. Odwoływane są wizyty u specjalistów. A pan? A pan jest zadowolony z siebie. Pan tutaj staje, jak gdyby nigdy nic, i powtarza te wszystkie kłamstwa, którymi raczył pan nas od 6 miesięcy. 10 dni temu mówił pan: Mamy 900 respiratorów. Kiedy pan kłamie - wtedy czy teraz? Chyba że dokonaliście nowych zakupów u kolejnego handlarza bronią, bo w tym jesteście dobrzy. Pan śmie mówić o ograniczeniu kontaktów społecznych. Drodzy państwo, to przecież pan premier Morawiecki mówił: Nie ma się czego bać, pandemii nie ma, spotykajcie się. To przecież rząd premiera Morawieckiego wysłał miliony SMS-ów do polskich seniorów. Tak. A potem? Potem już się nic dla was nie liczyło. Zamiast z pandemią pan walczy z prawdą, a prawda jest taka, że doszliśmy do ściany. To jest opinia lekarzy, dyrektorów szpitali, ratowników medycznych, ale pan zachowuje się tak, jak gdyby ich dramatyczne apele do pana nie docierały. Czas spojrzeć prawdzie w oczy. Wiecie państwo, jacy oni są pracowici?

To jest właśnie prawda o tym, jak walczycie z pandemią. W sobotę w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie 12 osób czekało na SOR, żeby znaleziono dla nich miejsca w szpitalach zakaźnych. A w tym samym czasie wasza tuba propagandowa mówiła o tym, że połowa miejsc jest wolna. Cytaty z rozmowy ratowników medycznych: W całej Warszawie nie ma wolnych izolatek. Możemy gdzieś dalej pojechać - nie wiem gdzie. Ja bym cię pokierowała, ale naprawdę nie mam gdzie, nie ma takiej opcji.

Do tego zmusiła ich wasza nieudolność i fatalne zarządzanie służbą zdrowia. I pan próbuje nam dzisiaj wmówić, że ci ludzie, którzy spędzają po kilkanaście godzin dziennie w kombinezonach, ratując ludzkie życie, nie mogąc iść do toalety, nie mogąc zjeść posiłku, że to ci ludzie za mało się angażują, że to oni kłamią? Dlaczego, zamiast wspierać pielęgniarki, salowe, ratowników medycznych, lekarzy staracie się właśnie na nich zrzucić odpowiedzialność za wasze błędy i zaniedbania? Dzisiaj też pan o nim mówił, chodzi o budowę szpitala polowego na Stadionie Narodowym. Tak, muszę to przyznać. Gdyby to było pół roku temu, może wtedy nie słyszelibyśmy o kierowcy karetki ratunkowej z Garwolina, który kiedyś jeździł na ratunek innym, a gdy sam zachorował na COVID, to zmarł, bo przez wiele godzin nie znajdowano dla niego miejsca w żadnym szpitalu. Gdyby pan podjął tę decyzję pół roku temu, to może nie słyszelibyśmy o pacjencie, który czekając w karetce na podjeździe szpitala, dostał udaru. I nawet nie można go było zbadać tomografem. Ale wy nadal utrzymujecie, że poradziliśmy sobie najlepiej we wszechświecie z walką z COVID-em. Przypominacie cały czas, jak tragiczna sytuacja była we Włoszech, gdzie lekarze musieli wybierać, którego pacjenta podłączyć do respiratora, a którego odłączyć, żeby zrobić miejsce innemu. Twierdzicie, że u nas tak nie jest? Stępińska mówi, że jest zamknięta, wysłali pismo. Nie mają personelu, nie przyjmują, a mi dusi się pacjentka.

I teraz, szanowni państwo - to nie będzie śmieszne, chociaż ten cytat brzmi groteskowo - zagadka dla pana: Przygotowałem plany na jesień. Teraz czas na wakacje.

Jak przygotował Polskę? Jaki był ten plan? Przeczytam panu rozdzierające serca słowa z mediów społecznościowych: Tata i dziadek chorowali na COVID. Dziadek zmarł w czwartek, tata w niedzielę. Tata chorował 3 tygodnie. Nikt, pomimo błagań, nie przyjechał taty zbadać. Nie chciano przysłać karetki, informowano mnie jedynie, że w szpitalach nie ma miejsc. Tata słabł, coraz trudniej oddychał, skarżył się na ból całego ciała. Mogłam mu towarzyszyć, stojąc pod balkonem, podając jedzenie i czekając na wynik. Tata zmarł w niedzielę.

Dziś prosicie nas o pomoc i przyznajecie, że kryzys was przerósł. Tak - mówię to z przykrością - nie daliście rady. Ale wiecie, dlaczego? Bo w czasach kryzysu potrzebni są odpowiedzialni politycy, którzy potrafią zarządzać gospodarką i służbą zdrowia. Tak, my umiemy to robić. Platforma Obywatelska i PSL przeprowadziły Polskę przez największy w historii kryzys gospodarczy. To wtedy, a nie teraz, panie premierze, Polska była stawiana za wzór. Ale wie pan, dlaczego? Bo wybraliśmy racjonalizm zamiast populizmu. Wiedzę ekspertów, a nie waszą strategię typu: jakoś to będzie. Odpowiedzialni politycy korzystają z wiedzy ekspertów, a nie z nimi walczą. Dzisiaj, gdy opinia publiczna widzi wasze zakłamanie, apelujecie do opozycji o współpracę. Pytam zatem: Gdzie byliście, gdy składaliśmy 16 dobrych projektów ustaw? Gdzie byliście, gdy składaliśmy 120 senackich poprawek? Gdzie byliście, kiedy chcieliśmy wspólnie pracować? Odpowiem panu, gdzie pan był. Pan zachęcał starszych ludzi do pójścia na wybory. Zachęcał pan, bagatelizując pandemię. Odrzuciliście każdą naszą inicjatywę, tylko dlatego, by doprowadzić do wyborów. Ale Polacy nie zasłużyli na to, by umierać z wami. Dlatego apeluję do pana: obudźcie się. To najwyższy czas, by spojrzeć na to, co dzieje się w Polsce, oczami zwykłego człowieka. Nie zza przyciemnianych szyb limuzyn, ale oczami tych najsłabszych, na autentyczny, realny świat, pełen ludzkich lęków i niepewności. Ten, który było słychać w tych tragicznych rozmowach, które przytoczyłem wcześniej. Tak, panie premierze, to czas, by zwrócić się do Polaków o solidarność, ale też powiedzieć o tym bardzo wyraźnie: Drodzy rodacy, ten rząd nie zdał egzaminu. Państwo ledwie dyszy podpięte do respiratora. Rządzący oblali ten egzamin, bo uznali, że można nie przejmować się ludzkim życiem, bo ministrowie pokazani arogancję, butę i krótkowzroczność. Bo handlowali maseczkami, bo zamawiali przepłacone respiratory. A później chcieli sobie zagwarantować bezkarność. Tak, panie premierze, ma pan dobre informacje, właśnie tutaj jest napisane, że taką dobrą szczepionką jest solidarność. Ale solidarność, którą należy dobrze rozumieć: to empatia, wzajemna pomoc, odpowiedzialność i samokontrola. Mam jeszcze taki apel, apel do was, Polacy: proszę, bądźmy wobec siebie życzliwi, dbajmy o siebie, dbajmy o innych.

Pomyślmy o innych. Wiem, że to jest niewygodne, ja też nie lubię nakazów czy zakazów, ale w trudnych czasach trzeba być solidarnym. Na koniec, panie premierze, tak Koalicja Obywatelska będzie współpracować z każdym, aby nieść pomoc Polakom. Ale nie zastąpimy rządów w działaniach, nie zastąpimy PiS w podejmowaniu decyzji. Wreszcie nie zastąpimy premiera Kaczyńskiego, który jest od 6 października odpowiedzialny za bezpieczeństwo, za zdrowie i życie Polaków. Możemy jednak podzielić się wiedzą i doświadczeniem. Tak teraz uczynię. Panie premierze, na pana ręce przekażę te 16 dobrych projektów ustaw, 120 poprawek. Przekazuję je panu, wierząc, że pan z nich wreszcie skorzysta. Tam jest zawartych pięć filarów walki z pandemią: 5 mld zł na walkę z epidemią, 100 tys. testów dziennie, 10 mln szczepionek na grypę, rzetelna informacja o stanie służby zdrowia. I dostęp do służby zdrowia dla pacjentów ze schorzeniami. Ale na Boga, panie premierze, wreszcie przeczytajcie te propozycje, choć raz posłuchajcie ekspertów samorządowców.

O głos poprosił pan premier Mateusz Morawiecki.

Wysoka Izbo!

To pierwsza sprawa. Drodzy Rodacy!

w czasach Platformy Obywatelskiej?

Dzisiaj to jest ok. 2 tys. więcej niż w waszych czasach. To się stało w ciągu 5 lat. Ile w czasach Platformy Obywatelskiej poświęcano środków na służbę zdrowia? Panie pośle Budka, panie przewodniczący, dziękuję za przypomnienie waszej strategii.

To była wasza strategia: likwidacja szpitali, komercjalizacja szpitali. Jak rządziła Platforma Obywatelska, zobaczcie, co się działo ze statystykami. Najlepiej, drodzy państwo, obrazuje to jedna zasadnicza liczba. Ile wydajemy na służbę zdrowia dzisiaj? Ile to było w czasach Platformy Obywatelskiej? Tyle mógłbym odpowiedzieć na te kłamstwa, które padły z tej mównicy, jak również na to, co mówił przewodniczący o jesiennej fali. Ale zakończę w ten sposób: sprostowałem kłamstwa, ale dalej wyciągam rękę.

Dlatego w naszej ustawie, którą dzisiaj tutaj wnosimy. A jest to któraś z kolei ustawa COVID-owa, któraś z kolei, która odpowiada na autentyczne potrzeby, a nie - w taki sposób przedstawiana rzeczywistość, jak to tutaj próbował pan przewodniczący Budka przedstawić. A więc, drodzy państwo, mimo wszystko, mimo tych kalumnii wyciągamy rękę do zgody. Czas na zgodę, dzisiaj jest czas na zgodę.

Dzisiaj jest czas na zgodę. Prosiłabym, żebyśmy jednak w tych wystąpieniach odnosili się do tematu dzisiejszego, żebyśmy rozmawiali o sytuacji dzisiejszej w służbie zdrowia. Bardzo dziękuję. Panie Premierze! czy ilość kłamstw na sekundę bije wszelkie rekordy.

Macie coś takiego jak GUS. I druga rzecz, pani marszałek, jeżeli chodzi o budowę szpitali. 33 szpitale mniej. 208 szpitali więcej. niech pan nie odwołuje prezesa GUS-u za te dane, okej? Chciałam bardzo wszystkich państwa poprosić o spokój. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Włodzimierza Czarzastego, klub parlamentarny Lewica. No spokoju to nie będzie. Wysoka Izbo! Szanowny Panie Premierze! Panie Jarosławie Kaczyński! Panie Mateuszu Morawiecki! Zwracam się do was obydwu, ponieważ nie wiem, który z was tak naprawdę rządzi.

Nie macie odpowiedzi, ale już wiecie, że to ważne. To zadam wam dzisiaj kilka pytań, żeby nie było, że nikt, panie premierze, o to nie pytał. Czy rząd wie, jak ma funkcjonować energetyka w Polsce, gdy załogi firm energetycznych zostaną zdziesiątkowane przez koronawirusa? Czy wiemy, kto zadba o to, aby do polskich domów płynął prąd? Czy rząd wie, kto dostarczy do polskich domów gaz, gdy zdziesiątkowani zostaną pracownicy w gazownictwie, w wodociągach? Czy rząd wie, kto zadba o dostawy żywności? Czy jesteście gotowi na najgorsze? Czy zrobiliście wszystko, do czego jesteście prawnie zobowiązani, abyśmy w naszym kraju mieli zapewnione zaopatrzenie w żywność i w wodę, bezpieczeństwo na drogach i na ulicach, ochronę przed napadami na nasze domy i mieszkania, zaopatrzenie w energię elektryczną, w gaz i inne surowce energetyczne, zaopatrzenie w takie paliwa, jak benzyna, olej napędowy, zaopatrzenie w ciepło systemowe i indywidualnie w węgiel; aby była ciągłość usług z zakresu łączności i sprawnych sieci teleinformatycznych; aby był dostęp do naszych pieniędzy i nieprzerwane usługi finansowe; aby pracowały usługi transportowe, w tym sprawne drogi i transport publiczny; aby funkcjonowały usługi komunalne, w tym odbiór odpadów, utrzymanie czystości w miastach; aby zapewnić ochronę przed spekulacją oraz w sytuacjach koniecznych stworzyć system reglamentacji produktów i usług koniecznych do życia; aby funkcjonowały usługi ratownicze; aby była ciągłość działania wszelkich służb państwowych, w tym Policji i administracji publicznej? Pewnie zdziwili się panowie premierzy, że odpowiadają osobiście i konstytucyjnie za tak wiele spraw i dziedzin, ale tak jest. Po prostu jesteście panowie za to odpowiedzialni. W związku z tym kolejne pytania. Czy posiadacie aktualny raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego? Nie posiadacie. Jak pan mówi, ja przez telefon nie odpowiadam. Jest taka zasada. Tata powinien nauczyć. Czy posiadacie uwzględniający pandemię narodowy program ochrony infrastruktury krytycznej? Czy zadbaliście o to, aby powstały wojewódzkie, powiatowe i gminne plany zarządzania kryzysowego? Nie zadbaliście. Pan na to pozwolił, panie Macierewicz, a pan się na tym zna. A przecież NIK stwierdził niedawno, że Polska nie ma skutecznego systemu ochrony ludności. Czy w ogóle wiecie, o czym mówię? Czy jako administracja podjęliście rozmowy i ustalenia z prywatnymi wytwórcami żywności, z właścicielami infrastruktury energetycznej, gazowej, transportowej i komunikacyjnej? Z dostawcami ciepła i wody, z sektorem finansowym?

Zadaję te pytania, choć praktycznie znam na nie odpowiedź. Ta odpowiedź brzmi: nie. Nie zrobiliście nic, abyśmy byli przygotowani na najgorsze.

Czy został przyjęty, panie premierze, panie premierze Kaczyński, panie premierze Morawiecki? Żeby nie było. Daję wam materiał do natychmiastowych przemyśleń, bo chcę wam pomóc. Nie będziecie musieli kraść naszych pomysłów. Czy jest państwowa strategia komunikacji ze społeczeństwem? Ludzie muszą wiedzieć, ludzie mają prawo wiedzieć, co ich czeka. Obudźcie się, bo w budynkach rządowych i w waszych mieszkaniach też może zgasnąć światło. Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Gawkowski, Lewica. Wysoka Izbo! Wysłuchaliśmy pana premiera i jak zwykle dowiedzieliśmy się, że jest dobrze.

Życzę, panie premierze, żeby pan miał taką werwę w walce z wirusem, z jaką pan tutaj odpowiada posłom i posłankom. W całym kraju brakuje łóżek, a wy mówicie, że się nic nie dzieje. Wczoraj w Krakowie pan Roman spędził 7 godzin w karetce, jeżdżąc od szpitala do szpitala. 83-letnia pani Barbara z Warszawy dowiedziała się, że na test może liczyć w piątek. Dziś jest środa. Nie ma sprzętu, a personel medyczny pracuje praktycznie bez snu. Umierają setki ludzi, nie tylko na COVID. Zapomnieliście o innych. Kazaliście odwołać operacje. Ludzie umierają, a wasi politycy mówią: tak musi być. To prawda. Śmierć nie wybiera, ale prawdą jest, że ludzie umierają przez was. Wszyscy przez ostatnie miesiące mówili, że obawiamy się scenariusza włoskiego. Tyle, że wy zafundowaliście Polakom scenariusz polski. Mieliście pół roku na to, żeby się przygotować. Nie robiliście nic. Zamiast pracować kłóciliście się, kto obsadzi więcej ministerstw. Przez 4 miesiące robiliście rekonstrukcję, bo pan Zbyszek pokłócił się z panem Mateuszem i trzeba było jakoś to pogodzić. Zachowywaliście się jak dzieci w piaskownicy. Utopiliście 70 mln w wyborach, które się nie odbyły. Sami nie pracowaliście, ale nie chcieliście też liczyć na innych. Lewica wielokrotnie dawała wam projekty. Z tej mównicy zgłosiliśmy ponad 1 tys. poprawek. Daliśmy wam plan „Bezpieczni przed drugą falą” Proponowaliśmy 100 tys. testów dziennie. Nie potrzeba. 2 mld na służbę zdrowia. A wy co? Oddaliście to na telewizję propagandową. Chcieliśmy szkoleń dla personelu, przekwalifikowania lekarzy. Słyszeliśmy - panikujecie. Dzisiaj pan premier powiedział: mamy ich sporo. Zobaczymy za 2 tygodnie. Ale po co? Jakoś sobie dadzą radę. Tutaj pan minister siedział do tej pory. Nie, wszystko w porządku. Czy pan się tego nie wstydzi? Czy pan naprawdę ma sumienie mówić Polakom, że jest tak dobrze? To dlaczego jest tak źle? Kiedy Polska stoi nad przepaścią, apelujecie o rozwagę. Pan dzisiaj z tej mównicy mówił o solidarności. Sami jesteście elitą i zbudowaliście tutaj państwo dla siebie. Wy nigdy nie będziecie spędzać czasu w kolejce po test. Wasza karetka zawsze będzie miała gdzie podjechać. W szpitalu zawsze będzie dla was łóżko i respirator. Wy nie znacie słowa solidarność, o którym pan tu mówił. Umiecie myśleć tylko o własnym interesie. Panie Premierze!

Czy pan wie, że zakażonych koronawirusem od początku jest ponad 1 tys. lekarzy, ponad 3 tys. pielęgniarek i położnych? Zamiast dziękować medykom za ich poświęcenie, próbujecie zrzucić na nich odpowiedzialność za swoje błędy i głupotę. Tacy jesteście. Chcecie wyjść z kryzysu, zwalając winę na innych, wczoraj na polityków opozycji, kilka dni temu na lekarzy. Zaraz powiecie, że to wina chorych. Tylko niech pan doda, że to może dlatego, że nie jedli jabłek. Ale to wy zawiedliście, nikt inny. To, że miliony polskich rodzin stracą członków rodzin, to wasza wina. To, że setki tysięcy tracą pracę i nie będą miały na czynsz, to również wasza wina. Za wasze błędy, za wasze zaniechania i waszą arogancję dziś płacą Polki i Polacy, ale kiedyś przyjdzie czas rozliczeń. Zostaniecie rozliczeni za wszystkie słowa, za nieodpowiedzialność, za brak strategii, za brak pomysłu, jak walczyć z koronawirusem. Rząd nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom i nie nadaje się do rządzenia. Rząd, który naraża zdrowie i życie swoich obywateli, powinien trafić pod sąd.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Żeby dobrze postawić diagnozę i wdrożyć leczenie, trzeba znać historię pacjenta, trzeba przebadać go fizykalnie, trzeba przeprowadzić wywiad. Jaka jest historia naszej walki jako państwa polskiego z koronawirusem? Rządzący w styczniu: epidemia jest bardzo daleko, w Chinach, może w ogóle do Polski nie dojść. W lutym: na wszystko jesteśmy przygotowani, na każdy scenariusz i wariant. W marcu: nikt się nie spodziewał takiej skali, nie spodziewaliśmy się, że ta epidemia nas tak dotknie. W maju już święcenie triumfu: najlepsi w Europie. W czerwcu: zwycięstwo nad koronawirusem. W wakacje: wirus w odwrocie, już jest mniej zjadliwy. We wrześniu kluczowe słowa Andrzeja Dudy: panujemy nad epidemią, epidemię mamy pod kontrolą. Utraciliście kontrolę nad państwem, utraciliście kontrolę nad epidemią. To jest akt oskarżenia wystawiany nie przez nas, polityków, nie przez opozycję. To jest akt oskarżenia wystawiany przez tysiące nowych zachorowań codziennie i setki zgonów. To jest akt oskarżenia, który będzie was gnębił każdego dnia. Jak dzisiaj jako opozycja, jako obywatele Rzeczypospolitej mamy zaufać słowom pana premiera? Pamiętam nawoływanie do współpracy w marcu. Na ten apel, wszyscy, jak tu jesteśmy, odpowiedzieliśmy pozytywnie. Uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach w kancelarii premiera, u prezydenta, z ministrami.

Wrzutka, o której nawet premier Emilewicz, bo z nią wtedy telefonicznie rozmawiałem, nie wiedziała. Żeby przejść dalej, dzisiaj zabrakło jednego słowa, panie premierze, kluczowego. Nie do nas, bo my jesteśmy politykami, możemy się tutaj spierać, dyskutować, ale do chorych, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracowników socjalnych, ekspedientek w sklepach, do całego społeczeństwa.

Słowa mogą zabijać, słowa mogą ranić, ale słowa, np. dla pacjenta, dają też nadzieję i przywracają życie.

Wtedy każda decyzja podejmowana była na wniosek prezydenta, wszystkie sztaby były pod jego nadzorem. Polska nie funkcjonowała bez mrugnięcia okiem pana prezydenta, a dzisiaj go nie ma. W ustawach, które wtedy wprowadziliście, było też wiele głupot. Za 70 mln na wybory można by było przebadać wszystkich mieszkańców Chodzieży, Andrychowa albo Aleksandrowa Łódzkiego. Mogliście nie wprowadzać restrykcyjnych zapisów wobec lekarzy. Z jednej strony mówicie „zaangażujmy się wszyscy” i dajecie takie przesłanie dla obywateli, a z drugiej strony wprowadzacie obostrzenia w Kodeksie karnym, które dają bezwzględne więzienie dla lekarzy, a bezkarność+ dla urzędników.

Jest 10 tys. zakażonych, są godziny w kolejkach do karetek, jest rozpacz pracowników medycznych, utrata zdrowia fizycznego i psychicznego, wyczerpanie w tym względzie.

Nie ma wprowadzonych tych rozwiązań, które by doceniały tak ciężko pracujących.

Jesteśmy gotowi do tej współpracy, tak jak cała opozycja dzisiaj zadeklarowała, dlatego że to jest wspólna odpowiedzialność, że nie wolno poświęcić na ołtarzu walki politycznej celu najważniejszego, jakim jest życie i zdrowie. Po pierwsze, w obszarze ochrony zdrowia: utrzymanie sprawności i wydolności szpitali. Szpitale, żeby ratować życie, muszą same żyć, muszą funkcjonować. Jeżeli one przestaną to robić, to wszystkie inne tarcze nigdy nie zadziałają. Dobrze, że o tym mówił pan minister Niedzielski. Ale my proponujemy coś innego. W prywatnych szpitalach, w prywatnych gabinetach - a tych miejsc jest 33 tys., ponad 400 szpitali, ponad 40 tys. gabinetów specjalistycznych - leczmy tych chorych, którzy cierpią na nowotwory, na choroby cywilizacyjne, na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, którzy chcą diagnostyki, leczenia w innych przypadkach, nie tylko w przypadku COVID-19.

Tych chorych nie wolno zostawić samych. Prywatne gabinety - otwarte za darmo, bo za nie ma zapłacić rząd.

Ale w sierpniu uważaliście, że tego nie będzie.

Bo to umożliwi zatrzymanie transmisji. My dzisiaj nie mamy jednego ogniska w Polsce. Nie jest tak jak po weselu w Nawojowej czy po wydarzeniach w kopalni. Dzisiaj ta transmisja jest niewidoczna i nie znamy miejsca i ognisk. To jest kolejny punkt. Podejście regionalne, rozmowa z samorządami, konsultacje i takie działanie, które nas nie wyznacza i nie nakazuje nam czegoś tylko i wyłącznie, ale też prosi o pomoc organizacje społeczne, fundacje. W gospodarce oczekujemy, domagamy się i żądamy zatrzymania wszystkich prac nad ustawami podnoszącymi podatki, wycofania się z ustawy, która wyprowadza ludzi na ulicę, bo są zdesperowani, bo stracą pracę, wycofania się z piątki przeciwko polskiemu rolnictwu. Niedziele handlowe powinny być przywrócone na czas epidemii, żeby chronić seniorów, żeby dać im szansę. Wreszcie napiszmy wspólny plan pandemiczny, bo jego po prostu brakuje. Rzucacie się od ściany do ściany. Najlepszym przykładem są maseczki. Jak chcecie przekonać pana Brauna i pana Bosaka, żeby nosili maseczki, skoro wasz minister zdrowia mówił, że one nic nie dają, że one nie chronią? Później mówił, że trzeba je nosić do wynalezienia szczepionki. Ale przyszedł przekaz z Nowogrodzkiej, że będą wybory - to trzeba nosić tylko jeszcze przez kilka dni, a później trzeba iść na wybory. Tu nie ma wiarygodności, nie ma strategii i nie ma spójności.

Moi Drodzy! Jeszcze jedna rzecz, apel już teraz nie do pana premiera, ale do episkopatu, do hierarchów Kościoła katolickiego. Zbliża się dzień Wszystkich Świętych, później Dzień Zaduszny. Dajcie jasny sygnał wiernym, że w tym roku lepiej poczekać, lepiej pójść kilka dni później, a nie dokładnie 1 czy 2 listopada.

Dzisiaj nie widzę siły w rządzących, żeby mogli samodzielnie tę kontrolę przywrócić. Dlatego zwracam się do moich rodaków: moi drodzy, szanowni państwo, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, dzisiaj my jesteśmy w stanie przywrócić kontrolę nad państwem, opanować sytuację swoją odpowiedzialnością, braterstwem, opieraniem swoich relacji i swoich poczynań na wiedzy, a nie na jakichś plotkach czy fake newsach.

Bardzo proszę, pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja.

Panie Premierze! Panie premierze, muszę powiedzieć, że zainspirował mnie pan, bo puścił pan nagranie pana Borysa Budki sprzed kilku miesięcy. Ja też mam tutaj takie nagranie. Od tego nagrania zaczniemy. Puszczam. Już większość osób tutaj, widzę, jest bez maseczek. Bo rzeczywiście cała ta choroba na szczęście została zwalczona, jest pod kontrolą, jest taka jak inne. Jest wiele różnych chorób, nie będziemy się ich bali na zapas, rząd wygrał z koronawirusem” Panie premierze, jesteście największymi hipokrytami i cynikami w historii polskiej polityki. A pan, panie premierze, jest na czele tego nierządu. Zamknęliście firmy, zamknęliście ludziom możliwości zarabiania pieniędzy, potem stworzyliście tarcze antykryzysowe. Tarcze antykryzysowe tworzyliście na bazie nie tego, że trwały jakieś konsultacje z przedsiębiorcami, tylko w ekipie, która tworzyła te tarcze antykryzysowe byli politycy PiS, którzy nie bazowali na swoich doświadczeniach, tylko na stwierdzeniu: wydaje nam się, że w ten sposób powinno się pomagać. Tysiące pracowników zostało zwolnionych albo ich pensje zostały obcięte lub zostali oni zmuszeni do podpisania aneksów dotyczących obniżki pensji do końca tego roku np. do 60%. Mówiliście, że narażacie całą gospodarkę, żeby kupić sobie czas. Chcieliście przez te 6 miesięcy przygotować nas na kolejną falę czy na to, co teraz się dzieje. No i jak przygotowaliście?

Zastanawialiście się tylko nad tym, jak zrobić rekonstrukcję rządu, kto będzie nowym ministrem czego. Wielka rekonstrukcja, wielka redukcja, redukcja, która skończyła się tym, że utworzyliście już trzy nowe urzędy i właściwie nic się tam wielkiego nie stało poza jakimś drobnym przemeblowaniem. Przez te pół roku nie potrafiliście nawet wprowadzić obostrzeń tak, żeby to było zgodne z prawem, przez co my to krytykujemy i negujemy. Skoro dzisiaj wprowadzacie tutaj prawo mówiące o tym, że maseczki będą musiały być noszone, no to znaczy, że wszystko, co działo się wcześniej, było bezprawiem. Anulujcie ludziom te mandaty, wtedy będzie to uczciwe. Chcę, żeby to wybrzmiało wyraźnie. To, co zrobiliście przez te lockdowny, to jest zbrodnia na polskiej gospodarce. To, co zrobiliście ludziom prowadzącym własne firmy, to jest niewybaczalny błąd, katastrofalny w skutkach. Mamy w tym momencie rekordowy w historii deficyt budżetowy. Mamy największy od 30 lat spadek PKB. Niestety tego się nie odrobi, dlatego że przeżeraliście lata, w których było dobrze. To jest coś, za co cały pana rząd i anonimowi doradcy, o których my się pytaliśmy, ale ich nazwisk niestety nie jesteśmy w stanie od pana uzyskać, będą musieli kiedyś zostać pociągnięci do odpowiedzialności przed sądami. Nigdy wam tego nie podarujemy. Polacy wam tego nie podarują, bo Polacy widzą, co się dzieje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja. Wysoki Sejmie! Panie Premierze! W pierwszych słowach swojego wystąpienia pragnę pozdrowić tych, którzy protestują w obronie swoich miejsc pracy, którzy próbują przetrwać w tym trudnym czasie epidemii i obostrzeń sanitarnych, ale także obostrzeń gospodarczych. Pragnę pozdrowić tu o rolników, którzy dzisiaj w całym kraju wychodzą, protestując przeciwko zabijaniu polskiej hodowli, zabijaniu polskiego eksportu, zabijaniu polskiego rolnictwa. Pragnę pozdrowić też branżę sportową, która liczyła na to, że zostanie potraktowana tak jak inne, i dziś traci nadzieję na to, że będzie mogła funkcjonować i przetrwać drugą falę epidemii.

Ci ludzie zasługują na to, żeby nazwy tych grup, które protestują i chcą przetrwać, padły z tej mównicy i żeby przypomnieć, że to, że polska gospodarka radzi sobie nie najgorzej, to nie jest zasługa pana premiera, to nie jest zasługa urzędników, to nie jest zasługa nawet tych, którzy wypłacają świadczenia z tarczy finansowej. To jest zasługa milionów ciężko pracujących Polaków i setek tysięcy ludzi prowadzących działalność gospodarczą, którzy codziennie myślą o tym, jak przetrwać ten trudny czas, a rząd rzuca im kłody pod nogi. W tych ustawach, które dziś wprowadzacie rzekomo po to, żeby ratować sytuację w ochronie zdrowia, która jest zawiniona przez wasze pięcioletnie zaniedbania, znów uderzacie w polskich przedsiębiorców. Wprowadzacie możliwość karania przedsiębiorców pod pretekstem łamania reżimu sanitarnego. Wystarczy jedna drobna (Dzwonek) kara, jeden drobny mandat za to, że ktoś nie założył maseczki, i pod znakiem zapytania stoi możliwość wydatkowania pieniędzy z tarczy finansowej. To jest skandal, co próbujecie przeforsować w tych przepisach, i nie pierwszy. Podobnie jest z wątpliwościami co do spółek komandytowych. Jeśli spółki komandytowe spróbują się przekształcać, to co z pomocą z tarczy finansowej? Pan Paweł Borys udzielił odpowiedzi, że nie będzie trzeba jej zwracać, ale to nie odpowiedź pana Pawła Borysa czy nawet komunikat PFR-u są wiążące. Dlatego apeluję w imieniu tych wszystkich, których dotykają wasze restrykcje: przestańcie im przeszkadzać i pozwólcie ludziom przetrwać ten kryzys, a zajmijcie się tym co ważne, czyli ochroną zdrowia. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę, pani poseł Hanna Gill-Piątek, poseł niezrzeszony. Wysoka Izbo! Panie Premierze! Panie Ministrze! Ponieważ padło tutaj dzisiaj bardzo wiele słów o solidarności, chcę skupić się na jednym bardzo konkretnym problemie. Chcę z tej mównicy być głosem tych, których zazwyczaj się nie słyszy, czyli głosem ponad 30 tys. osób bezdomnych, które w tym systemie w tej chwili, podczas epidemii muszą jakoś się zmieścić. Nie mieszczą się.

Te schroniska i noclegownie funkcjonowały w trybie zamkniętym podczas epidemii wiosną, ale teraz, w tym momencie bardzo wiele osób, które żyje poza nimi, zgłasza się. Bardzo wielu bezdomnych szuka schronienia w schroniskach i noclegowniach. I powstaje problem, kto ma płacić za ich testy, kto ma organizować im kwarantannę. Bo jedna osoba zakażona w schronisku, które liczy 150 podopiecznych, naprawdę może spowodować taką katastrofę, z jaką mamy do czynienia bardzo często w domach pomocy społecznej. Dobrym przykładem jest Gdańsk, który nie czekając na to, aż się ustali kompetencje, kto ma realizować ten obowiązek, już faktycznie zbudował kontenery na czasową izolację. I tam to funkcjonuje bardzo dobrze, ale to jest inicjatywa samorządu.

Natomiast ja podniosłam telefon i zadzwoniłam do NFZ-u, zapytałam co mogę zrobić, żeby zrobić bezpłatny test tak dostępny osobie nieubezpieczonej. I wiecie państwo, co usłyszałam? Że muszę iść do lekarza pierwszego kontaktu, ponieważ osoba nieubezpieczona musi być ubezpieczona, żeby taki test zrobić. A więc dla bezdomnego te testy tak naprawdę są niedostępne. Chciałam zapytać w takim razie, co rząd zrobi, żeby ludzie podczas pandemii, ludzie bezdomni, nie zamarzali tej zimy na ulicach. Bo ten problem trzeba bardzo pilnie rozwiązać i organizacje prowadzące schroniska i noclegownie bardzo czekają na to rozwiązanie. Dziękuję.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Warto tutaj kilka tych nieprawd i kłamstw sprostować. Otóż raporty GUS-u, na które powoływał się pan przewodniczący Borys Budka, jasno mówią o tym, że w 2012 r. zmieniliście statystykę i zamieniliście filie na szpitale. Czyli coś, co nie było szpitalem wcześniej, [[Oklaski]] nagle się stało szpitalem. To tylko dlatego pan przewodniczący mógł tutaj zacytować coś takiego. Mało tego, z raportu GUS, uwaga: Z uwagi na zmiany prawne - ustawa o działalności leczniczej - mające wpływ na sposób wyodrębniania i rejestracji placówek, w tym szpitali, dane dotyczące liczby szpitali są nieporównywalne z danymi z lat poprzednich. Liczba szpitali odnosi się do przedsiębiorstw albo wydzielonych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne. sprostowanie.

To partia, która nie troszczyła się o słabszych, dla której programy społeczne, dla której dbanie o słabszych ludzi. o ludzi leczonych w szpitalach w godny sposób nie miało znaczenia. Przypominam strategię Arłukowicza, który mówił do wojewody właśnie o tym, żeby zamknąć cztery szpitale. Jak jeszcze można to uzasadnić i udowodnić? No, w bardzo prosty sposób. Właśnie poprzez to, że zajmowaliście się tylko i wyłącznie tymi. Poziom środków przeznaczonych na służbę zdrowia bardzo wyraźnie to podkreśla. I dlatego dzisiaj w takiej dziwnej koalicji Konfederacja i Koalicja Obywatelska, Konfederacja i Platforma Obywatelska razem, nagle. I jedni poprzez ignorowanie tego, jak groźna jest dla naszej gospodarki ta pandemia, i drudzy, którzy dążą do zamknięcia natychmiastowego wszystkiego, są poważnym niebezpieczeństwem dla naszego państwa, poważnym niebezpieczeństwem dla całej polskiej gospodarki. A teraz moje słowa. Szanowni państwo, proszę zobaczyć, spojrzeć na wykres spadku zakażeń w czerwcu i przypomnieć sobie, czego wszyscy wtedy chcieliśmy. Chcieliśmy otwierania gospodarki, wzrostu handlu, handlu międzynarodowego, usług. I właśnie wtedy trzeba było walczyć o gospodarkę, dbać o gospodarkę, bo ile, jak długo, 2, 3 miesiące gospodarka może być całkowicie przymrożona? Wiadomo, że nie. Dlatego pod koniec czerwca, w lipcu, tak jak dbaliśmy o powrót normalnych usług leczniczych, szpitalnych, o czym mówił pan minister Niedzielski, tak samo dbaliśmy o to, żeby w III kwartale gospodarka polska ruszyła z powrotem z kopyta. Tak się zresztą stało.

Teraz pan poseł Dziambor - niestety pomylił się, mówiąc o deficycie najwyższym.

Dzisiaj na skutek wzrostu gospodarczego jest to daleko mniej. Drodzy Rodacy! Tym, którzy straszą co do stanu gospodarki, chcę powiedzieć, opowiedzieć - może tak powinienem powiedzieć - jedną ciekawostkę. Otóż w ostatnim czasie udaje nam się plasować obligacje na rynkach z rentownościami ujemnymi, a to oznacza wzrost gospodarczej wiarygodności Polski na rynkach międzynarodowych. Nie ma lepszego sposobu sprawdzenia wiarygodności niż „głosowanie” przez różne podmioty międzynarodowe i krajowe swoimi własnymi środkami na emisje obligacji, które nigdy nie były w taki sposób wyceniane na rynkach międzynarodowych, tak dobrze dla nas. To świadczy o tym, jak świat patrzy na nasz rozwój gospodarczy. Teraz mowa o lockdownie. Drodzy państwo, tak jak powiedziałem, musimy nauczyć się żyć, pracować, kształcić bez lockdownu całkowitego, choć nie wiadomo, jakie decyzje trzeba będzie podejmować. Wczoraj czytam o Irlandii, która mówi o tym, że trzeba zrobić niemal całkowity lockdown, w niektórych obszarach głębszy niż wiosną. To dlatego rozbudowujemy bazę łóżkową, rozbudowujemy liczbę szpitali - nie tych fikcyjnych, statystycznych, o których mówił pan przewodniczący Budka, tylko tych faktycznych. Nie ma już pana przewodniczącego Czarzastego, ale chcę też powiedzieć, że i te sformułowania były zupełnie nieprawdziwe. A poza tym proszę nie zwracać się do nas per „wy” bo to jest zwyczaj z poprzedniej epoki, z PRL-u, a dzisiaj żyjemy w wolnym kraju. Szanowni Państwo!

Drodzy rodacy, nie tylko nie przeczę, ale z najwyższą dozą współczucia i szacunku wobec wszystkich tych, którzy w obecnym stanie rozwoju epidemii doświadczają problemów, krzywd, o których słychać, o których wiemy, że są. Wiadomo, że wszystko, co robimy, ma usprawniać funkcjonowanie całego systemu służby zdrowia. Szpitale nie podlegają państwu.

Dlatego dziękuję medykom. Proszę również wszystkich o to, żeby byli jak najbliżej pacjentów. Jednocześnie odpowiadam panu przewodniczącemu czy panu prezesowi Kosiniakowi-Kamyszowi, który mówił o premiowaniu bądź niepremiowaniu.

Nasze dane, które porównujecie państwo z danymi z Unii Europejskiej, potwierdzają, że do tej pory ta równowaga, droga środka sprawdza się lepiej niż w wielu innych przypadkach.

Wysoka Izbo! To nie jest pana najlepszy dzień. Kilka konkretnych liczb. Rok 2020 - spadek o 20 tys. O 20 tys. zmniejszyliście liczbę łóżek szpitalnych. Są jeszcze gorsze dane.

Pan przeszkadza dzisiaj przez cały dzień. Bardzo dziękuję. Panie Premierze! Pan dobrze zauważył, że nasz projekt dotyczy wszystkich lekarzy - 1500 zł dla lekarzy, pielęgniarek, wszystkich medyków i pracowników społecznych - a wasz projekt dotyczy tylko tych, których skieruje do pracy wojewoda. To nie jest tylko i wyłącznie. One są kosztowne - 900 mln miesięcznie - ale to jest wynagrodzenie dla tych, którzy pracują na pierwszej linii frontu. Wy w swojej ustawie mówicie o tych, których skierujecie do pracy, a my mówimy o tych, którzy pracują od marca.

Wysoka Izbo! Panie Premierze!

Elita. Brak solidarności. To najmniejszy z zarzutów, które powinniśmy wam dzisiaj stawiać. Narzekacie, że my dzielimy. Panie premierze, w tamtym tygodniu we wtorek, nie tak dawno, na spotkaniu z panem przedłożyłem cztery projekty ustaw. Pan powiedział: będziemy rozmawiali. Chciałem zapytać, panie premierze, co z trzema pozostałymi? Pomożemy przedsiębiorcom w czerwonych strefach? A może pomożemy ludziom, którzy tracą pracę?

Minister zdrowia już w marcu wydał polecenie do Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym ten dodatek został określony dokładnie na tym samym poziomie, jaki jest w przypadku lekarzy skierowanych do walki z COVID-em. A teraz, jak tylko ustawa ewentualnie po przegłosowaniu wejdzie i 200-procentowe wynagrodzenie ustali, to oczywiście minister zdrowia wyda odpowiednie polecenie Narodowemu Funduszowi Zdrowia, żeby płacił też medykom zatrudnionym. I tutaj też chciałbym to powiedzieć. Właśnie onkologia, o której mówił pan Kosiniak-Kamysz, jest również taką dziedziną, którą. Przez całe wakacje, co podkreślałem w moim wystąpieniu, staraliśmy się utrzymać ciągłość i stabilność pracy onkologii.

To jest pewna wyspa, której chcemy pilnować ze względu na priorytet polityki rządu. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do pytań.

Jako pierwszy pan poseł Tomasz Latos. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Właściwie należałoby zacząć od prostowania tych wszystkich innych danych, które były przytaczane. Ja tylko powiem chociażby o jednej liczbie. Panie przewodniczący, w roku 2015 w ratownictwie medycznym funkcjonował na polskim rynku podmiot zagraniczny. Państwo nieraz się musieliście wcześniej tłumaczyć z różnego rodzaju braku koordynacji między Państwowym Ratownictwem Medycznym a tym prywatnym. To tyle, jeżeli chodzi o historię. Natomiast, panie premierze, panie ministrze, bardzo dobre, rzeczowe wystąpienie, bardzo gratuluję. Myślę, że warto jeszcze powiedzieć o danych dotyczących chociażby tych dodatkowych szpitali, które będą tworzone. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Premierze! Od marca wiemy, że pandemia jest w naszym kraju, a dzisiaj bardzo dużo czasu w tych wystąpieniach poświęca pan historii tego, co było 5, 6, 10 lat temu. Ja liczyłam, że z pana dzisiejszego wystąpienia dowiem się, jak rząd wykorzystał ten czas i co zrobił, żebym mogła obywatelom powiedzieć, co ich czeka, jakie są procedury. Przypominam, że jak mówiłam na początku o tym, że pojawia się pandemia, słyszałam, że straszę Polaków. Potem słyszałam, że dobrze, że był początek w innych krajach, bo my się do tego lepiej w Polsce przygotujemy. Dzisiejsze wystąpienie pana premiera i żadnej dobrej informacji dla Polaków.

I to jest realny problem Polaków. Pani poseł Katarzyna Kotula, klub Lewicy. Panie Marszałku! Panie Ministrze! No tak, faktycznie. Zabraliście 34 geriatryczne łóżka ze Szpitala Wolskiego w Warszawie, a teraz chcecie odbierać łóżka pacjentów ze Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Jedne i drugie zostały ufundowane przez WOŚP - WOŚP, który w okresie totalnej zapaści psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej zakupił 798 łóżek i obdarował nimi 34 oddziały w Polsce. Panie Premierze! Panie Ministrze! Mam pytanie: Komu jeszcze odbierzecie łóżka szpitalne, jakiego rodzaju pacjentów pozbawicie stosownego leczenia, bo zamiast zajmować się planowaniem strategii walki z pandemią i przygotowaniem planu na drugą falę, zajmowaliście się walką o stołki i łagodzeniem wewnętrznych konfliktów, wciskając w tym czasie obywatelom kit o tym, jak to nie jesteście dobrze przygotowani? Dlaczego nie zaplanowaliście odpowiednio wcześniej zamówień, zakupów medycznych. szczególnie że cały sprzęt zakupiony przez WOŚP jest wyprodukowany w Polsce, jest dostępny w polskich fabrykach? Bardzo proszę. Pani poseł, pani skończyła już wystąpienie, proszę opuścić mównicę. Pani poseł, czy pani rozumie, co ja do pani mówię? Ale jak dokończyć? Jest minuta albo nie ma.

Panie Ministrze Zdrowia! Lekarz rezydent pyta, ilu pielęgniarzy, lekarzy, pielęgniarek, lekarek przeszkoliliście do obsługi pacjentów COVID-owych i sprzętu COVID-owego od marca tego roku.

To są poważne zagrożenia, na które nie reagujecie. I co za zły wam podpowiedział, żeby w tym trudnym czasie koronawirusa wprowadzać tzw. piątkę Kaczyńskiego, ustawę wprowadzającą embargo na polskich rolników, na polskie rolnictwo, i od miesiąca wyciągać ich do Warszawy, na drogi, gdzie naprawdę nie da się zachować warunków kwarantanny, warunków izolacji?

Przed przyjściem do Sejmu powiedział pan w mediach, że te przepisy z tej kolejnej specustawy są niezbędne do walki z wirusem. To proszę powiedzieć: Co was powstrzymywało do tej pory przed wprowadzeniem tych przepisów? Ogłosił pan, że w Katowicach szpital będzie tworzony w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a przecież w Katowicach jest wolny szpital przy ul. Ceglanej, który jest niezakontraktowany, stoi pusty, do wzięcia od zaraz. Dlaczego zapychacie szpitale ludźmi z łagodnymi objawami, podczas kiedy oni tego naprawdę nie potrzebują, i potem jęczycie, że nie macie miejsc w szpitalach? Jeśli będziecie przyjmować tylko tych, którzy naprawdę potrzebują opieki, to skończy się problem z dostępnością miejsc w szpitalach. Pan poseł Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość. Też nie ma? Pan poseł Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Po wysłuchaniu tej informacji właściwie można zadać tylko jedno pytanie: Czy pan celowo okłamuje Polaków, czy pan naprawdę tak niczego nie wie i niczego nie kontroluje? Naprawdę pan wierzy w te słowa, które pan mówi? Wymienia pan tutaj liczby: 2 tys. respiratorów wolnych, 45% obłożenia, jeżeli chodzi o te, które są wysłane do szpitali, a ludzie umierają, bo nie mogą się doczekać na respirator. To pan chce powiedzieć, że pan trzyma w magazynach respiratory, a nie daje pan ich ludziom, żeby nie umierali? To chce pan powiedzieć? Pan dzisiaj się chwali liczbą testów, że 60 tys. to tak dużo? Przecież to jest ułamek, ułamek tego, co robią cywilizowane kraje. Pan zdaje sobie sprawę, że te 60 tys. to jest tyle, ile duże miasta europejskie robią na swoje potrzeby? Zdaje pan sobie z tego sprawę? Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Główne ogniska koronawirusa są w dużych miastach. Jednak z powodu pandemii cierpią również mieszkańcy wsi, w tym wielu rolników. Stąd moje pytanie: Ilu rolników i członków ich rodzin zostało od początku pandemii skierowanych na kwarantannę? W jaki sposób państwo udzieliło im pomocy, aby mogli kontynuować swoją produkcję? Dotyczy to przede wszystkim produkcji zwierzęcej, która wymaga codziennej troski o zwierzęta. Drugie pytanie dotyczy wielkich zakładów produkujących żywność. W ostatnich tygodniach ognisko COVID-19 wykryto w zakładach mięsnych w miejscowości Ujeździec Mały koło Trzebnicy, w Suwałkach, w Szczecinie i w Starachowicach. Stąd moje drugie pytanie: Czy rząd ma plany na zapewnienie Polakom dostaw żywności w sytuacji, gdy na kwarantannę będę kierowane załogi największych zakładów produkujących żywność?

Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sporo uwagi w swoim wystąpieniu, zwłaszcza na początku, poświęcił pan współpracy, solidarności, wspólnemu stawaniu przed tym wyzwaniem, jakim jest pandemia.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Rozpocznę od podziękowań.

Ja przypomnę państwu, że z państwa strony, Platformy Obywatelskiej, prominentna polityk mówiła o tym, że starszym ludziom nie warto wszczepiać stawu biodrowego, bo i tak się nie wyrehabilitują, a do lekarza chodzą dla rozrywki. Dziękuję za to, że mamy najniższy wskaźnik zgonów z powodu COVID-u. A przypomnę, że wszystkie rankingi mówią, że to we Francji, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii rzekomo są wspaniałe systemy ochrony zdrowia, tymczasem Polska ma najniższy wskaźnik umieralności z powodu COVID.

Uważnie słuchałem pana, panie premierze, i można odnieść wrażenie, że pan już w ogóle nie walczy z tą epidemią. W ogóle tylko tworzy pan dla siebie alibi.

Proszę zwrócić uwagę, jak pan mówił dzisiaj. Przecież pan w ogóle nie walczył z epidemią. Pan walczył z Platformą, dzisiaj walczył pan z panem Budką, wczoraj walczył pan z panem Giertychem. Bo pan ma walczyć z COVID-em jako polski premier, a nie z opozycją, a nie z adwokatami, politykami czy z parlamentarzystami. Pan mówił o milionach szczepionek, które pan ma. To co pan powie tym ludziom w aptekach, którzy się odbijają od aptek, którzy codziennie słyszą: nie ma szczepionek? Lewicy.

Panie Premierze! Rząd wprowadził dla nich pewne uprawnienia, ale one istnieją niemal tylko na papierze. I tutaj przytoczę kilka przykładów. Teleporady - świetny pomysł idący z duchem czasu, ale nie działa. Albo nie można się dodzwonić do lekarza, albo nawet jak można, to i tak w większości przypadków trzeba przyjść z dokumentacją medyczną. Dofinansowanie szczepionki na grypę - doskonale, tylko nie ma tych szczepionek. Ani w przychodniach, ani w aptekach, ani w hurtowniach. Starsi ludzie często godzinami stoją przed przychodnią, żeby dostać się do lekarza, ryzykując zarażenie. Puszczają im nerwy. Były przypadki, że konieczna była interwencja Policji. To nie koniec. Seniorzy mają problem nawet z podstawowymi sprawami w pandemii. Obowiązek noszenia maseczek nie jest dofinansowany przez państwo, a maseczki jednorazowe kosztują nawet złotówkę. Miesięcznie to jest kilkadziesiąt złotych, co naprawdę przy ogólnej mizerii polskich emerytur stanowi duży wydatek.

Bardzo proszę, pani poseł.

Niech pani zada pytanie. przekłamań dotyczących kwalifikacji personelu pielęgniarskiego.

Pan poseł Dariusz Joński, klub Koalicja Obywatelska. Jeszcze nie. Panie Marszałku! Zadaję dość proste pytanie: Kiedy będzie strategia, tak aby ludzie nie umierali? Tak jak ten ratownik medyczny, kierowca pogotowia, który został zarażony koronawirusem, jeździł od szpitala do szpitala na Mazowszu. Co pan zrobi, kiedy będzie strategia, aby dyspozytorka nie musiała płakać, tak jak dzisiaj w szpitalu w Poznaniu, kiedy musiała powiedzieć, że nie ma wolnego miejsca? Może będzie za godzinę, kiedy niestety ktoś umrze. Kiedy w końcu będzie strategia, abyście nie kupowali od handlarza bronią respiratorów i testów z Korei, które nawet w Korei są nieużywane? A polskie szpitale odsyłają. Kiedy w końcu wyjaśnicie, dlaczego siłownie i baseny, a nie kościoły i kluby taneczne? Gdzie w tym wszystkim logika? Pani poseł Joanna Borowiak, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Premierze! Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że posłowie opozycji nawet w sytuacji epidemii, kiedy walczymy z wirusem, nie potrafią odstąpić od politycznej walki. Dzisiaj też liderzy opozycji pokazali i próbowali mówić z tej mównicy tak, by zrealizować swoje polityczne cele. Słuchając opozycji, jestem wdzięczna za to, że w Polsce nie rządzi dziś Platforma z koalicjantami. Bo dziś kazaliby nam, tak jak w czasie epidemii świńskiej grypy w 2010 r., cieszyć się wiosną, spać i pracować spokojnie, kiedy Polacy umierali. Albo powtarzaliby za swoim politycznym guru, że to nie epidemia, a histeria globalna. Nie dbaliście o służbę zdrowia, o ochronę zdrowia. Nie potrafiliście myśleć perspektywicznie. Dlatego dzisiaj, choć teraz, od tego momentu, posłuchajcie apelu pana premiera Morawieckiego.

Panie Premierze! Ten obraz obiegł całą Polskę. Dziś co pan proponuje?

Ile to będzie kosztowało? Ile z tego tytułu przybędzie miejsc pracy? Kto panu doradza? Czy pan nie pamięta, że 31 lipca 2019 r. powołał pan pełnomocnika rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego w randze wicepremiera, dzisiaj funkcjonującego? Powołał pan 2 lata wcześniej Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Czy pan o tym nie pamięta? Czy nie należy tych ludzi zdyscyplinować, a pieniądze na dodatkowe miejsca pracy swoich kolesiów przeznaczyć na nowe miejsca, na nowe łóżka? Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! Dziękuję za to dzisiejsze wystąpienie, za jasną informację, ale przede wszystkim dziękuję za pracę służb, wojewodów, sanepidu i wszystkich, którzy starają się w tym trudnym okresie pomagać, w odróżnieniu od opozycji. Ja w odróżnieniu od opozycji nie mam kontaktu, nie mam informacji tylko z Internetu, bo jestem na bieżąco w kontakcie z tymi, którzy się chorymi zajmują. Zarówno z dyrektorem mojego szpitala, jak i panem wojewodą. Panie Premierze! Sytuacja w Małopolsce jest naprawdę trudna, o czym pan dobrze wie. Dobrze, że mamy sprawnego wojewodę.

Wniosek o dodatkowe środki, który wpłynął wczoraj, wczoraj też dotarł do pana. Jestem w kontakcie. Mam nadzieję, że ta pomoc. Panie Marszałku! Panie Premierze! Zmarnowaliście 6 miesięcy i zostawiliście Polskę bezbronną. Nie zrobiliście nic, aby przygotować nas na drugą falę epidemii, za to bawiliście się jak na Titanicu, wydając setki milionów złotych, kiedy te pieniądze były potrzebne chorym. Ale w jednym jesteście mistrzami: w zaklinaniu rzeczywistości. Te wasze zapewnienia, że sytuacja jest pod kontrolą, że dajecie radę, że cały świat nas podziwia i nam zazdrości. Dziś w świetle codziennych danych o zmarłych i zakażonych te wasze zaklęcia nie są śmieszne, są zwyczajnie żałosne. Jestem z Małopolski, gdzie sytuacja jest wyjątkowo dramatyczna. Brakuje lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych. A co robi PiS-owska władza?

Panie Premierze!

Odpowiedział na szereg waszych wcześniejszych spostrzeżeń, co było działaniem rządu w wakacje, co było działaniem rządu w ostatnich tygodniach, co będzie strategią na najbliższe lata. Dlaczego nie jesteście w stanie nawet potwierdzić, że jest strategia i są działania rządu?

Wysoka Izbo! Dzisiaj mamy do czynienia z poważnym pożarem, którym jest oczywiście epidemia, ale także sytuacja w ochronie zdrowia. Igraliście z żywiołem, igraliście z ogniem i teraz pali nam się dom, cały system przestaje być wydolny. Jako opozycja chcemy wam pomóc, chcemy was wspierać w tych działaniach, w tych wszystkich zadaniach. Podamy wam wodę, nie podamy wam wiadra z benzyną, jak to jest nam często sugerowane i zarzucane, ale to pan, panie premierze, musi być dzisiaj strażakiem, który gasi pożar, a nie go wznieca. Zatem proszę o ugaszenie pożaru w szpitalu wojewódzkim w Sosnowcu, gdzie brakuje podstawowego sprzętu, gdzie brakuje podstawowych lekarstw, gdzie za chwilę przestanie istnieć oddział toksykologii. To jest poważny problem, panie premierze, a to wszystko w wyniku wojenki wewnętrznej w PiS. Pan poseł Konrad Frysztak, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wyjaśnię, przybliżę panu to, z czym borykają się Polacy niebędący Kaczyńskim, Sasinem czy Czarnkiem. Co pan powie tym, którzy wczoraj przez 7 godzin stali w jedynym punkcie poboru wymazów w Radomiu, punkcie dla Radomia i powiatu radomskiego?

Dziś, panie premierze, to samorządy, te znienawidzone przez was samorządy, przepraszam, przez wasze ugrupowanie, walczą za was z koronawirusem. To szpitale powiatowe, te, które zamykaliście, walczą z koronawirusem. To one dziś toczą walkę. Panie pośle, pan już skończył.

Szanowny Panie Premierze! To jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Może czas skończyć z tym teatrem pozoru i propagandy? Koronawirus nie wybiera. Rząd się wyleczy, ale Polacy niekoniecznie, dlatego zadaję pytanie: Dlaczego nie chcecie chronić Polaków? Szczepienia na grypę. Zalecenia Unii Europejskiej: 75% populacji. Francuzi, Włosi szczepią 75% populacji, Polska - 4%.

Dlatego przytoczę panu słowa: Ludzkie nieszczęścia po drodze będą bolesną nauką dla rządu. Bardzo proszę, pan minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szanowni Państwo! Odsiewając deklaracje od rzeczywiście zadanych pytań, bo większość z tych wypowiedzi miała charakter deklaracji politycznej, chciałbym zacząć od tematu łóżek. Jeżeli chodzi o łóżka, proszę pamiętać, że Polska jest krajem, który w porównaniach międzynarodowych ma zdecydowanie największą liczbę łóżek w przeliczeniu na 100 tys. obywateli. My w tych statystykach wyprzedzamy wszystkie kraje rozwinięte, wszystkie kraje Europy Zachodniej, i to wyprzedzamy w sposób bardzo znaczący.

Druga informacja jest taka, że jeżeli patrzymy na średnie poziomy zajętości tych łóżek w poszczególnych latach, to widzimy, że w roku 2019 ten poziom zajętości wynosił 66%, czyli 2/3. To jest taka wielkość, która wydaje się stabilna. To, co robimy, zmieniając model służby zdrowia czy ochrony zdrowia w Polsce w ostatnich latach, to jest stopniowe przenoszenie ciężaru lecznictwa z poziomu szpitalnego na poziom ambulatoryjny, czyli zamieniamy pobyty wielodniowe, które były związane chociażby z diagnostyką, które trwały wiele, wiele dni, w szpitalu, na takie intensywne jednodniowe procedury diagnostyczne.

To tak naprawdę był zabieg, który urealnił tę liczbę.

Wcześniej prowadzący szpitale czy inne podmioty lecznicze wpisywali do rejestrów prowadzonych u wojewodów tę liczbę bez żadnych konsekwencji, czyli mogli deklarować dowolnie dużo, a właśnie pojawił się weryfikator tej liczby, bo trzeba było to zapełnić personelem. W wyniku wprowadzenia tych norm odbyła się tak naprawdę akcja budowania pewnej większej przejrzystości i wiarygodności danych. To jest efektywne przedsięwzięcie, które polega na tym, że urealniliśmy tę liczbę łóżek - do tych, które mają obsadę, które nie są papierowymi łóżkami w żaden sposób niereprezentującymi realnej wartości.

Tak naprawdę dyskusja o tym jest powodem do oddzielnej debaty, do oddzielnej informacji. Szczepionki.

Proszę pamiętać, że producenci szczepionek planują dostawy na rynek w oparciu o to, co miało miejsce w zeszłym roku.

Do końca października to będzie 240 tys. To są już podpisane i zakontraktowane szczepienia. W listopadzie mamy największą dostawę, ponieważ to jest optymalny czas na szczepienie. Kumulacja grypy w zeszłym roku miała miejsce na przełomie stycznia i lutego, a najlepsza odporność po szczepionce jest mniej więcej do 60 dni. Jeżeli chodzi o grudzień, tutaj też przewidujemy dostawę 200 tys. szczepionek. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o wydawanie respiratorów, to Ministerstwo Zdrowia tutaj bardzo ściśle współpracuje z Agencją Rezerw Materiałowych. Weryfikujemy, czy jest realne zapotrzebowanie na respiratory.

I mamy do czynienia z taką sytuacją, że w wyniku zapotrzebowania. Wydaliśmy w ciągu ostatnich 2 tygodni 700 respiratorów. Tak naprawdę non stop prowadzimy dialog ze szpitalami, szczególnie tymi właśnie, które są obciążane zadaniami COVID-owymi, po to, żeby te wielkości urealniać.

Te 60 jednostek podlega w tej chwili działaniom kontrolnym Narodowego Funduszu Zdrowia, który, jak wiemy, nie jest łatwym partnerem w trakcie kontroli.

Bardzo dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeszcze kilka odpowiedzi, refleksji, które tutaj padły, w odpowiedzi na to, co zostało zgłoszone. I chyba taka kwestia, której dzisiaj nie omawialiśmy, a ona jest fundamentalnie ważna dla całego systemu, mianowicie: lekarze i kształcenie lekarzy. Otóż chcę podziękować z tego miejsca byłemu ministrowi zdrowia panu Konstantemu Radziwiłłowi za to. za decyzje, które zostały podjęte na samym początku naszych rządów, w 2016 r. Otóż wtedy zaczęliśmy kształcić o 50% więcej lekarzy. Drodzy państwo, drodzy rodacy, wiemy doskonale, ile czasu zabiera kształcenie lekarza: 6 lat - studia, potem 8–10 lat - specjalizacje. Wiemy doskonale, jak bardzo potrzebni nam są nowi lekarze. Jedną z pierwszych decyzji, które podjął dzisiejszy wojewoda, a ówczesny minister zdrowia, było zwiększenie naboru na studia medyczne.

Ale trzeba dobrze wiedzieć, kto rozpoczął ten proces, kto zajął się rzeczywiście tym bardzo żmudnym, długotrwałym problemem, tak żeby w strategiczny sposób ten brak nadrobić. Padały tutaj oskarżenia i oszczerstwa w kierunku poprzedniego ministra zdrowia dotyczące respiratorów.

Jeszcze raz dziękuję panu ministrowi Szumowskiemu, że przewidując drugą falę, rzeczywiście nabywał te respiratory już w maju, czerwcu i lipcu. Szanowni Państwo!

To tylko tak tytułem informacji, bo dzisiaj pielęgniarki anestezjologiczne czy przeszkalani interniści są bardzo ważni w kontekście całego procesu leczenia COVID-19. Co do tych punktów wymazów, o które tutaj były pytania, to chcę też powiedzieć, że oprócz tradycyjnych punktów wymazów tworzymy, już jest tworzonych, już funkcjonuje ponad 300 punktów wymazów, które też będą w coraz większym stopniu obsługiwane przez Wojska Obrony Terytorialnej i wojska operacyjne. Dlaczego? Po to, żeby pielęgniarki czy czasami inni medycy, którzy obsługują te punkty wymazów, mogli być uwolnieni do czynności medycznych, do czynności bardziej potrzebnych w służbie zdrowia w tym momencie. W ramach naszej trzeciej i czwartej linii obrony następuje już przesunięcie tych zasobów. Jednocześnie też dziękuję panu ministrowi obrony narodowej za to, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy, letnich miesięcy, nie czekając na rozwój wydarzeń, zaordynował przeszkolenie 100 tys. żołnierzy w zakresie właśnie kursów i szkoleń medycznych. Teraz są wśród nich ratownicy, którzy wchodzą w miejsca, które mogą być zwolnione przez medyków. Tak, jest Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, spotykamy się codziennie od wiosny. Wiosną spotykaliśmy się codziennie, potem latem zmniejszyliśmy częstotliwość, dzisiaj znowu spotykamy się codziennie. Jest tam zawsze sprawozdanie ministrów dotyczące spraw dzisiaj najważniejszych, tego, ile jest łóżek, ile jest respiratorów (Dzwonek), jak sprawić, żeby było ich jeszcze więcej, jak lepiej zapewnić dystrybucję. Tak, mogę tylko raz jeszcze zaapelować do wszystkich samorządowców, bo to oni często są organem założycielskim. Jeżeli potrzebujecie respiratorów, to są one dostępne. Jeżeli potrzeba zmian organizacyjnych, proszę się... jeżeli potrzeba jakiegoś sprzętu.

Była mowa też o karetkach. Przybyło kilkaset karetek w ciągu ostatnich 2 lat, a więc to usprzętowienie służby zdrowia. Myślę, że jak spytacie większość dyrektorów szpitali, to potwierdzą, że nigdy nie było takiego zastrzyku finansowego i zastrzyku w zakresie sprzętu dla szpitali.

Otóż wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, żeby się porozumiewać z samorządowcami, żeby niektóre szpitale były przekształcane w szpitale COVID-owe. Na tym ten proces dzisiaj polega. Uzgadniamy z samorządowcami, które szpitale jakie usługi medyczne mają świadczyć. Dziękuję za głos dotyczący bezdomnych. Przyjrzymy się temu, jak wygląda leczenie osób bezdomnych czy zgłaszanie się przez osoby bezdomne na testy. Szanowni Państwo! Chcę tylko raz jeszcze na koniec podkreślić, że dziękuję za pozytywne głosy. Czas na zgodę. Jesteśmy gotowi do pozytywnego, konstruktywnego dialogu.

Do wynalezienia szczepionki, lekarstwa, tego oczywiście dokładnie nie wiemy. Ale niezwykle ważne jest to, żeby w zgodzie była cała klasa polityczna, bo to dzisiaj jest test, nie tylko dla rządzących, dla rządzących absolutnie też.

Chcę z całą mocą podkreślić: odrzucamy skrajności, odrzucamy tych, którzy nie chcą stosować rygorów i będziemy bezwzględnie egzekwować poprzez nasze służby mundurowe wszystkie te obostrzenia i rygory. wszystkie usługi, wszystkie branże. Nie najwyższą w Polsce, ale dmuchamy na zimne. Chcemy te niezłe parametry gospodarcze utrzymać, bo praca, praca i jeszcze raz praca dla Polaków jest najważniejsza. Będziemy o to dbać, równocześnie i równolegle z walką z COVID-19. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie informacji.